Sejm propozycję przyjął. Ten sprzeciw przegłosujemy. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła w dyskusji w pierwszym czytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydium Sejmu proponuje, aby w dyskusjach nad pozostałymi punktami porządku dziennego Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

Kto się wstrzymał?

Sejm propozycję przyjął. Proszę. Szczęść Boże! Rok temu w jednym z warszawskich szpitali dziecięcych zmarł chłopczyk, Szymonek, zostawiony na śmierć przez nieludzkich ludzi. Już nie tylko dzieci nieurodzone nie są w Polsce bezpieczne, ale także te, które się urodziły zdrowe, nie mogą liczyć na opiekę i gwarancję bezpieczeństwa ze strony państwa polskiego.

Proszę bardzo, pan poseł Krzysztof Gawkowski, Lewica, wniosek formalny. 1 minuta, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

O szpitalach jednoimiennych mówimy od kilku tygodni. Sytuacja, która tam panuje, jest po prostu dramatyczna. Personel najzwyczajniej na świecie panikuje. Nie wiedzą, co robić, nie mogą z nikim porozmawiać, a ministerstwo nie chce pomagać. Mówimy też o pacjentach, którzy jeszcze bardziej to odczuwają, bo zdają sobie sprawę, że dzisiaj szpitalne jednoimienne, dedykowane do walki z pandemią, są pozostawione same sobie. Pandemia jest elementem, który cały czas rośnie.

Nie, to nie jest wniosek formalny. Bardzo proszę, z wnioskiem formalnym, panie pośle.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Szanowni Państwo! Ta sprawa musi być wyjaśniona i potrzebna jest w tym zakresie informacja premiera. Jak to się stało, Wysoka Izbo, że w Ministerstwie Zdrowia pojawił się handlarz bronią? Jak to się stało, że bez żadnego trybu, przy autoryzacji służb państwa PiS, podpisano umowę na 250 mln zł bez określenia tego sprzętu? Jak to się stało, że z 12 tys. respiratorów zamówionych za 44 mln zł nie dostarczono żadnego respiratora?

To nie jest wniosek formalny, panie pośle. Naprawdę. Przyjmę go, ale to nie jest wniosek formalny. Ale dziękuję panu bardzo.

Proszę podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej panią Annę Surówkę-Pasek o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Szanowna Pani Marszałek! Szanowne Panie, Szanowni Panowie Posłowie! Jest to projekt, który realizuje zapowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy, które dotyczyły wsparcia polskich rodzin w wypoczynku, zwłaszcza tym wakacyjnym, a także wsparcia branży turystycznej. Pierwszym z nich jest wsparcie rodzin. Świadczenie w postaci bonu turystycznego, którego wartość wyniesie 500 zł, będzie przysługiwało wszystkim tym rodzinom, które pobierają świadczenie 500+, a także tym rodzinom, które mają dzieci w pieczy zastępczej i z tego tytułu otrzymują stosowne świadczenia. Ważne jest również to, że rodziny, które opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, będą mogły uzyskać prawo do dodatkowego bonu. Oznacza to, że rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym na jedno dziecko będą mogły uzyskać łącznie kwotę 1000 zł, co, jak ma nadzieję pan prezydent, pozwoli na zorganizowanie wypoczynku nie tylko takiemu dziecku, ale także opiekunowi, który z tym dzieckiem będzie mógł spędzić czas.

Żeby dzieci, które później nabędą prawo do tych świadczeń, miały również możliwość skorzystania z tego bonu, ten bon będzie można wykorzystać do końca marca 2022 r. Co jest bardzo ważne, wartość tego bonu jest zwolniona z podatku dochodowego, ale także nie będzie wliczana do wysokości dochodu, od którego zależy nabycie prawa do różnego rodzaju świadczeń. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, dlatego że nie wpłynie ono na dotychczasowe świadczenia, które będzie pobierała rodzina. Warto również zauważyć, że ten bon będzie można wykorzystać wielokrotnie, aż do momentu wyczerpania się kwoty, na którą on opiewa. Ewentualna kontrola, czy ktoś ma prawo, czy nie do takiego świadczenia, będzie miała charakter następczy.

To jest drugi cel tego projektu ustawy, wsparcie polskiej branży turystycznej, albowiem bon ten będzie można wykorzystać u przedsiębiorców turystycznych, a także w organizacjach pożytku publicznego organizujących różnego rodzaju wyjazdy czy imprezy turystyczne, działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Branża turystyczna, jak wiadomo, w wyniku COVID-19 dość mocno ucierpiała. Niedawno byłam na śniadaniu prasowym, w którym uczestniczyli przedstawiciele branży turystycznej. Są oni bardzo zadowoleni z propozycji wprowadzenia takiego instrumentu, który niewątpliwie posłuży do zminimalizowania negatywnych skutków związanych z pandemią, a także z przestojem, który nastąpił na skutek zamknięcia różnego rodzaju obiektów turystycznych. Wysoka Izbo!

Bardzo dziękuję, pani minister. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwsza, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, głos zabierze pani poseł Urszula Rusecka. Pani Minister! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko wobec przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym z druku nr 423. Szanowni Państwo! Prezydencki projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym jest wynikiem zapowiadanego już w kwietniu programu wsparcia polskich rodzin z jednej strony, a pomocy branży turystycznej z drugiej.

Sprawnego przywódcę poznajemy po tym, jak radzi sobie nie wtedy, kiedy jest dobrze, ale w czasie kryzysu. Od kilku miesięcy świat zmaga się z potężnym kryzysem zdrowotnym wywołanym epidemią i będącym jej następstwem kryzysem ekonomicznym. Tylko dzięki ogromnemu wysiłkowi oraz dobrej współpracy rządu Zjednoczonej Prawicy i prezydenta Andrzeja Dudy udaje się Polskę bezpiecznie przeprowadzić przez światowy kryzys. Świadczą o tym zarówno twarde dane, jak i opinie niezależnych światowych ekspertów z dziedziny ekonomii. I tak dla przykładu: na łamach niemieckiego portalu Focus Online czytamy, że Polska stała się fenomenem dla europejskich ekonomistów. Głównym czynnikiem decydującym o znaczącym ograniczeniu strat gospodarczych związanych z wirusem SARS-CoV-2 była szybka reakcja polskiego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości. Duży pakiet pomocowy uchronił polskie firmy od bankructwa i poważnej utraty miejsc pracy. Wysoka Izbo! Prezydent Andrzej Duda wraz z rządem Zjednoczonej Prawicy poprzez przełomowe społeczne i solidarnościowe programy inwestuje w polskie rodziny i w polski biznes, wzmacnia tym samym krajową gospodarkę. Wprowadzone rozwiązania spowodowały zwiększenie popytu wewnętrznego i dzięki nim polska gospodarka jest mniej podatna na zagrożenia i światowy kryzys. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów i może wyjść z pandemii wzmocniona - czytamy w „Die Welt” Pokonujemy kryzys zdrowotny. Dzięki działaniom rządu, ministra zdrowia polscy lekarze nie musieli i nie muszą wybierać, którego z pacjentów podłączyć do respiratora. Pokonujemy także kryzys gospodarczy. Dzięki kolejnym odsłonom tarczy kryzysowej i tarczy finansowej służącym wsparciu przedsiębiorców i ochronie miejsc pracy na chwilę obecną ponad 85 mld trafiło na konta polskich przedsiębiorców. Ochroniliśmy miliony miejsc pracy. Szanowni Państwo! Ustawa o bonie turystycznym autorstwa pana prezydenta Andrzeja Dudy to kolejny instrument wsparcia dla polskiej branży turystycznej i rodzin z dziećmi. Panie Prezydencie!

Jesteśmy przekonani, że będzie nam dane realizować wspólnie jeszcze wiele takich dobrych projektów dla polskich rodzin. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie opiniuje przedstawiony przez prezydenta projekt ustawy. Dziękuję.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie!

Nie wiemy, jak będzie wyglądać kondycja firm turystycznych na jesieni, kiedy skończy się przyjęte przez parlament w pierwszej tarczy tzw. odroczenie płatności za zaliczki, które klienci wpłacili na poczet niezrealizowanych imprez turystycznych.

W ostatnim czasie ze środowiska rządzących wyszedł projekt obliczony według mnie na efekt kampanijny, niedobrze rozpoznający potrzeby branży turystycznej dziś, tu i teraz.

Dziękuję za konsultacje wszystkim oprócz pana przewodniczącego, pana marszałka Terleckiego, który otrzymał ten projekt, ale nie zechciał się z nami spotkać, porozmawiać. Chcieliśmy to rozwiązywać ponad podziałami, bo gospodarka w takim kryzysowym czasie wymaga działania ponad podziałami.

To też pokazuje. Oczywiście w jakiś sposób ten projekt prezydencki zawiera pewien element wsparcia dla rodziny, tego nie będę jakby nie podkreślał, natomiast progospodarczym instrumentem nie jest i wyklucza bardzo wiele grup społecznych, które dla turystyki polskiej w takim kryzysowym okresie miałyby znaczenie.

To jest projekt progospodarczy. Panie pośle Suski, niech pan to przeczyta i zrozumie.

Pan o tym nie wie, że 60 mld, ponad 60 mld to jest wielkość sektora gospodarczego, którym jest turystyka. Pan chce jakimś wycinkiem działania, który ma być tylko ratunkiem, a według mnie się nie da uratować prezydenta Dudy, prezydenta Dudy w kampanii, za pieniądze publiczne. To jest.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rzeczywiście dzisiaj debatujemy nad projektem dotyczącym Polskiego Bonu Turystycznego i pewnie nie jest to przypadek, że dzieje się to na tydzień przed wyborami prezydenckimi. Nie jest to przypadek, bo zawsze, gdy widzę pana ministra i panią minister, wiem, że na pewno jakiś projekt prezydencki pojawia się w polskim parlamencie. I nie jest to przypadek, że pojawia się właśnie dzisiaj. I można powiedzieć tak: rzeczywiście dobrze się stało, że 10 maja te wybory się nie odbyły, bo gdyby się odbyły, to pewnie dzisiaj tego projektu byśmy w ogóle nie mieli w planie obrad polskiego parlamentu. Bo prawda jest taka, że jeżeli chodzi o branżę turystyczną, doskonale polski rząd wiedział, jakie ma ona problemy, już od początku marca br., w momencie kiedy zapadały decyzje dotyczące zamykania granic, zamykania hoteli czy zamykania w ogóle m.in. całej branży turystycznej. Doskonale wiedziano, że te problemy będą bardzo poważne, jeżeli chodzi o branżę, która - zwracam uwagę na jedną rzecz i myślę, że rządzący może z tego wyciągną wnioski - jest branżą zajmującą się nie tylko kwestią dotyczącą wynajmu miejsc w hotelach czy wynajmu bazy turystycznej. Przecież dzisiaj, i to mówią badania, złotówka wydana na turystykę generuje dodatkowe 4,3 zł w innych branżach, bo przecież turystyka to jest wzrost handlu, turystyka to jest wzrost wpływów, jeżeli chodzi o transport, turystyka to również wzrost wpływów, jeżeli chodzi o rolnictwo, turystyka to wzrost wpływów, jeżeli chodzi o inne dziedziny gospodarki.

Klub Lewicy w tej sprawie będzie składał stosowne poprawki. Trzeba się niewątpliwie zastanowić nad tym, czy rzeczywiście ten projekt ma dotyczyć tylko rodzin, które pobierają 500+, czy nie powinno się poszerzyć bazy osób, którym ten bon turystyczny będzie przysługiwał, chociażby o emerytów i rencistów. To jest bardzo istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju branży, bo prawda jest taka, że 40% wszystkich zamówień, jeżeli chodzi o noclegi, to są lipiec i sierpień, natomiast jest pytanie, co robić w pozostałych miesiącach.

Dziękuję. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pani Premier! Szanowni Panowie! Jak miało być, pani premier? Miało być szumnie zapowiedziane 1000 zł. Pieniądze miały trafić do 7 mln Polaków zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

Program miał obowiązywać 2 lata, budżet miał sfinansować 90%, przedsiębiorcy mieli sfinansować 10%.

Pytali rolnicy, pytali ci, którzy zrezygnowali z pracy, żeby się zajmować swoimi niepełnosprawnymi dziećmi lub też członkami rodzin. Była to pewna propozycja, która odpowiadała częściowo na to, co się dzisiaj dzieje, szanowni państwo, w branży turystycznej. A jaką mamy rzeczywistość? Wystarczy tylko zapytać, szanowni państwo, tych, którzy prowadzą restauracje, hotele. Zresztą sami chodzimy, widzimy, co jest. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. I ta propozycja, która była zaproponowana przez panią premier, była na pewno propozycją o wiele ciekawszą niż ta, nad którą dzisiaj procedujemy podczas tego posiedzenia, szanowni państwo.

Im się nic nie należy? Szanowni państwo, klub Koalicji Polskiej będzie miał dalej idącą propozycję i poprawkę, żebyśmy już przestali wreszcie na tej sali dzielić Polaków.

Muszę powiedzieć, szanowni państwo, co dobrego jest w tym projekcie, bo o tym też muszę powiedzieć. To, że on ma obowiązywać 2 lata - dobrze. To, że ma obowiązywać na terenie Polski - dobrze. To, że wyciągnęliście państwo wnioski, że ma to być w formie elektronicznej, cyfrowej - dobrze. To, że będzie ułatwiony sposób - okej.

Niestety zarówno senatorowie z PiS-u, jak i senatorowie z Platformy powiedzieli: nie, nie pomagamy tej branży, nie rozszerzamy im możliwości.

Zaproponowaliśmy już przy pierwszej tarczy fundusz płynnościowy. Dlaczego tyle miejsc pracy straciliśmy od tego czasu? Dlaczego dzisiaj, kiedy kończy się czerwiec, nie ma propozycji, żeby przedłużyć niektóre rozwiązania? Niektóre branże jeszcze przez wiele tygodni nie będą mogły funkcjonować. Państwo to widzicie. Dzisiaj polscy przedsiębiorcy tego oczekują. I my jako klub Koalicji Polskiej zgłosimy tę poprawkę, o której mówiłem, szanowni państwo.

Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!

Będziemy więc finansować tylko tę część społeczeństwa, która w waszym mniemaniu jeździ. Dlaczego nie dla wszystkich? Dlatego że przecież w tym projekcie nie chodzi o ratowanie żadnej turystyki. Wam chodzi o to, żeby dosypać, dać kolejne 500+ elektoratowi, który mógłby przypadkiem już zapomnieć, że 4 lata temu dostał od was te 500+, które już było, bo już się przyzwyczaił. Jest to standard, że ludzie się przyzwyczajają do pewnego dobra, które jest.

To nie jest prawda, ponieważ nie tylko wy to poparliście. To 500+ jest tak naprawdę pobraniem podatków w bardzo wysokiej kwocie, a potem oddaniem części, ponieważ jesteśmy tacy dobrzy. A wystarczyło odpodatkować Polaków. Jeżeli ten projekt, który teraz państwo próbujecie wprowadzić, jest wprowadzany dla ratowania turystyki, to dlaczego nie odpodatkować po prostu przedsiębiorców w branży turystycznej? Dlaczego nawet nie dać im 500 zł, choćby jako ulgę podatkową, jeżeli tak koniecznie chcecie się trzymać tych okrągłych liczb?

Przypisaliście to dzieciom, ponieważ jaką bestią trzeba być, żeby nie dać dzieciom na wakacje, żeby nie dać dzieciom, żeby przeżyły wakacje w tym ciężkim czasie koronawirusowym. Uratujmy dzieci. To jest szantaż, to jest szantaż reszty parlamentu, ponieważ ci, którzy zagłosują przeciwko, będą wytykani palcami jako ci, którzy nie dali dzieciom. Konfederacja temu szantażowi się nie podda. Powinniście odpodatkować Polaków w koronawirusie, tak jak mówiliśmy, a tego nie zrobiliście. I teraz też powinniście odpodatkować branżę turystyczną, czego nie chcecie zrobić, bo za to nie można sobie przypisać zasługi, tak jak za 500+ przelewem. Dziękuję bardzo. Z jednej strony dzieci - a dlaczego nie na każdy PESEL? Dlaczego po prostu nie zwiększenie kwoty wolnej od podatku? My takie rzeczy możemy z wielkim bólem serca zaakceptować, traktując to po prostu jako zwrot nadpłaconych podatków, które państwo bez litości ściągacie. Ale tu ukryty jest jeszcze po drugiej stronie tego równania pewien oszukańczy trik. Państwo chcecie, żeby ten bon był do realizacji poprzez, uwaga, przedsiębiorcę turystycznego. Prosty człowiek, nawet prosty poseł - nie każdy się doczyta, że np. hotelarz to już nie jest przedsiębiorca turystyczny. A zatem nie można ze swoim bonem elektronicznym pojechać tam, dokąd się chce, trzeba dać zarobić pośrednikom w tej branży, biurom turystycznym, które bardzo popieramy, i w ogóle bardzo nam się podoba to, że Polacy łebscy, zaradni, globtroterzy jeżdżą we wszystkie strony świata, dopóki ich władza nie zamknie we własnym kraju, ale. Pani poseł na pewno będzie miała czas, pan marszałek udostępni, prawda? Proszę tutaj, na trybunę, i proszę merytorycznie polemizować. Właściwie Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno się pochylić nad każdym projektem ustawy, który tutaj przepychacie w ostatnich tygodniach, miesiącach, bo to jest korupcja.

Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Sylwester Tułajew, klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi za tę kolejną inicjatywę ustawodawczą, kolejną, bo 33.

Za ten projekt chciałbym bardzo serdecznie podziękować, a także za tę aktywność. Czyny, nie słowa. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku dodatku solidarnościowego, tak teraz po raz kolejny prezydent pokazuje wiarygodność, pokazuje aktywność i po raz kolejny prezydent Andrzej Duda mówi: czyny, nie słowa.

Wysoka Izbo! Gdyby Sejm za rządów PiS był sercem demokracji, był miejscem prawdziwej debaty, dziś procedowalibyśmy tutaj, na tej sali, dwa projekty: pierwszy, wniesiony 9 czerwca przez klub Koalicji Obywatelskiej, projekt o bonie turystycznym, i drugi, który właśnie teraz procedujemy, który ujrzał światło dzienne wczoraj o godz. 14. Sezon turystyczny rozpoczął się majówką. Wiemy, że była pusta. Wakacje też nie będą takie, jak dawniej. Są to straty nie do odrobienia. Dziś procedujemy projekt, który dzieli ludzi, który dzieli Polaków, dlatego jako klub Koalicji Obywatelskiej będziemy starali się włożyć wszystkie te dobre poprawki z naszego projektu, który nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych, który wpisuje się w program nowej solidarności, który da realne wsparcie (Dzwonek), tak by stał się projektem, inwestycją, która. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani premier bardzo mocno walczyła o przejęcie w ramach umowy koalicyjnej od ministra sportu turystyki. Dostała turystykę. Cztery tarcze kryzysowe przewidują oczywiście rozwiązania dla branży, ale specjalnie jej dedykowanych tam nie ma. Czekano.

Dziękuję.

Wysoka Izbo!

Kiedy patrzę na inicjatywy pana prezydenta, to chciałoby się rzec, że mamy do czynienia z nową pięciolatką, pięciolatką w 3 dni, bo tyle jest nowych inicjatyw.

Postulowałbym, aby te środki były przyznane każdemu, kto chce wybrać się na zasłużony wypoczynek. Poseł Robert Winnicki, koło Konfederacja. Poseł Andrzej Gawron, klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Szanowni Państwo! Pandemia stawia bardzo duże wyzwania przed gospodarką, przed państwem, dotyczące tego, żeby tę gospodarkę uratować. Inicjatywa prezydenta absolutnie wpisuje się właśnie w to, że pomagamy przedsiębiorcom, pomagamy polskim rodzinom, pomagamy też osobom z niepełnosprawnościami. To jest też bardzo ważny punkt tego programu, ponieważ pomagamy najsłabszym. Szanowni Państwo! Myślę, że trzeba się zastanowić nad poszerzeniem zakresu firm, które w tym uczestniczą. O tym była mowa.

Panie Marszałku! Pani Premier! Później zmieniliście zdanie: nie wszyscy, tylko ci zarabiający do 5200 brutto.

Wpuszczacie w gospodarkę 3 mld zł i mówicie, że to ma uratować branżę. Tymczasem, po pierwsze, ten bon będzie realizowany przez 2 lata, w związku z czym duża część środków trafi do przedsiębiorców, jak już nie będą im potrzebne, a to w tej chwili jest najgorzej. Po trzecie, w Krakowie turyści rocznie wydają 6 mld zł. W związku z tym te 3,5 mld na 2 lata na całą Polskę to jest kropla w morzu potrzeb. Traktujecie przedsiębiorców niestety niepoważnie. Jeżeli chcecie pomóc firmom turystycznym, to musicie przedłużyć działanie tarczy pomocowej na kolejne miesiące, komunikować swoje decyzje wcześniej, a nie w ten sposób, że otwieracie granice i 3 dni wcześniej branża się dowiaduje (Dzwonek), że nagle może działać. Pan poseł Stefan Krajewski, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Otóż są polskie rodziny, które niestety czują się oszukane przez pana prezydenta i przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo jeszcze w maju obiecano im, że dostaną po 1 tys. zł w postaci bonu turystycznego na jedną pracującą osobę. Dzisiaj dla polskiej wielopokoleniowej rodziny, składającej się często z dwójki dorosłych, rodziców, emerytów, rencistów i dwójki pracujących dzieci, oznaczałoby to 4 tys. zł na wspólne, rodzinne wakacje. Tymczasem za sprawą jakichś wyborczych gierek te rodziny zamiast 4 tys. zł nie dostaną ani złotówki, a inne rodziny, zwane przez rząd statystycznymi, z dwójką małych dzieci dostaną na wakacje tylko 1 tys. zł, a miało być 4. Emeryci i renciści pytają, dlaczego nie dostaną ani złotówki. Branża turystyczna z województwa kujawsko-pomorskiego, z którego pochodzę, liczyła na te środki.

Wysoka Izbo! Czy my musimy stosować ciągle półśrodki? Teletombola, bony. Kiedyś były modne talony na małego fiata, dzisiaj bony rozdaje pan prezydent, rząd. A wystarczyłoby, żeby pan prezydent spełnił swoje obietnice wyborcze z 2015 r. Kwota wolna od podatku. Chociażby to w dużej mierze byłoby pomocą dla rodziców, dzieci. Chociażby kwestia wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców. To zostaje na lata. Z bonów wszystkich rozliczycie, bo z jednej strony jest pomoc z PFR, a z drugiej strony wzrosną dochody przedsiębiorców i już nie będzie 75%, tylko 50 albo 25.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Premier! Państwo Ministrowie! Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z rządem Zjednoczonej Prawicy zawsze wychodzi naprzeciw polskim rodzinom, polskim firmom. Szczególnie w czasie pandemii doskonale to widzimy. Państwo wiedzą, że największe problemy w obecnej sytuacji ma branża turystyczna. Dziękuję panu prezydentowi jako wnioskodawcy za tak wspaniały pomysł, jakim jest bon turystyczny. Do pani minister mam pytanie: Czy bon turystyczny nie będzie objęty opodatkowaniem i zostanie [[Dzwonek]] wyłączony z jakichkolwiek roszczeń egzekucyjnych?

Wysoka Izbo! Zmieńcie nazwę ustawy. To nie bon turystyczny, tylko obiecanki cacanki+. Od początku kluczycie. Najpierw chcieliście wykluczyć osoby na umowach śmieciowych, ale na szczęście, na skutek wywieranej przez nas presji, zmieniliście ten skandaliczny zapis, za to wprowadziliście wykluczenie rodzin bezdzietnych.

Karmicie nas pięknymi kłamstwami, a prawda jest taka, że nie stać was na to. I zobaczycie, że za chwilę przy urnach wyborczych Polacy powiedzą wam: mamy dość.

Panie Marszałku! Chciałam zapytać o długą listę przypadków, z którymi mamy do czynienia w kolejnych kampaniach. 500+ na drugie dziecko zostało wprowadzone w kampanii wyborczej. To samo z programem 300+. To wszystko państwa zdaniem przypadki? Tak wam po prostu wyszło, bez związku z kampanią? Nie jest to przekupywanie ludzi? Tym razem to zasługa wspaniałomyślnego prezydenta Dudy, który ma za wszelką cenę wygrać i pokornie kontynuować swoją misję notariusza w pięknym pałacu. Dalej chcecie wmawiać, że to nie jest projekt skrojony pod kampanię wyborczą? Jaką mamy gwarancję, zwłaszcza jeśli przegracie, że nie wycofacie się z tej propozycji? Oby z obietnic nie zostało okrągłe zero. Pani Premier! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję, że ten program jest.

Macie dość bycia w opozycji, bo nie stworzyliście żadnego przełomowego programu, tylko powtarzacie i plagiatujecie nasze programy. Jak mówiliśmy: 500+, to mówiliście: A dlaczego nie na każde dziecko? Jak daliśmy na każde dziecko, to: budżet się rozsypie. Wszystkim rozdajmy, ograniczmy podatki. No to życzę szczęścia. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest odpowiedzialnym rządem, odpowiedzialnym za budżet i za sytuację polskich rodzin. Tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości [[Dzwonek]] realnie przeprowadzi nas przez ten kryzys. Panie Marszałku! Szanowni Państwo Ministrowie! Chciałem zapytać: Dlaczego, prowadząc swoją kampanię wyborczą, pan prezydent nie wykorzysta tej okazji do tego, żeby rzeczywiście realnie pomóc branży hotelarskiej oraz sektorowi spotkań i konferencji? To one przecież ucierpiały najbardziej na skutek rządowych działań, bezprecedensowego ograniczenia praw obywatelskich.

Potrzebna jest sektorowa polityka, sektorowa tarcza w celu wsparcia przemysłu turystycznego, w tym branż spotkań i konferencji. Dziękuję. Pani poseł Anna Paluch, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.

To jest ważny projekt, który pomoże firmom turystycznym przetrwać.

I czy państwo nie wiecie, że przedsiębiorstwa turystyczne to są mikro-, małe, średnie i może większe przedsiębiorstwa, które mogą zgodnie z przepisami korzystać z tarcz, z kolejnych wersji tarczy antykryzysowej? Hotele, kwatery turystyczne mogą korzystać z rozwiązań, które tutaj omawiamy.

Panie i Panowie Posłowie! Panie Marszałku! 22 maja klub Koalicji Obywatelskiej rozesłał do wszystkich klubów w parlamencie projekt ustawy o bonie turystycznym. Czy działalność rolnicza, czy działalność gospodarcza - wszystkie osoby, które pracują, które dokładają się, można powiedzieć, do budżetu państwa, miały otrzymać bon w wysokości 500 zł, nawet, tak jak w tym projekcie, w postaci elektronicznej. Cieszy nas, że państwo czerpią inspiracje z naszych projektów. Jest to dla nas dobry sygnał, szczególnie że głównym celem bonu turystycznego było to, żeby wspomóc polskie przedsiębiorstwa turystyczne. Natomiast rodzi się kilka pytań. Dlaczego tak wybiórczo? Przecież tak naprawdę, realnie rzecz biorąc, obejmie to bardzo małą liczbę rodzin, ponieważ np. osoby z małym dzieckiem, które jadą do dziadków na wakacje, nie dostaną żadnych pieniędzy, a przede wszystkim nie dostaną ich studenci (Dzwonek), nie dostanie ich też bardzo wiele osób, które pracują i znowu nic nie dostaną od państwa. Wysoka Izbo! Od posłów PiS słyszymy tutaj o wielkiej odpowiedzialności ze strony rządu, pana prezydenta, w związku z tym projektem ustawy, nad którym dzisiaj procedujemy. To nie jest wyraz odpowiedzialności, a wręcz przeciwnie. Czy odpowiedzialne jest to, że państwo na początku obiecywaliście Polakom po 1 tys. zł, a dajecie 500 zł, i to nie wszystkim?

Mówimy o tym, że powinno być dla wszystkich tak samo. To po pierwsze. A po drugie, proszę państwa, patrząc na to, co państwo proponujecie, chcę wam powiedzieć, że Polacy są bardzo rozczarowani państwa propozycją, zarówno obywatele, jak i branża turystyczna, ponieważ nie odpowiada to na ich potrzeby.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To jest projekt na potrzeby kampanii wyborczej. Gdyby nie było dzisiaj kampanii wyborczej, najprawdopodobniej tego projektu by nie było. Ten projekt znowu dzieli. Czy panu prezydentowi nie zależy na emerytach, na rencistach, na osobach niepełnosprawnych czy na tych, które nie mają dzieci, ale bardzo ciężko dzisiaj pracują i ledwo wiążą koniec z końcem? Proszę państwa, skoro wszyscy wiemy, że branża turystyczna jest w bardzo trudnej sytuacji, to niech rząd wykorzysta jeszcze jeden element, ten, który jest do dyspozycji, czyli tzw. politykę fiskalną.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Piotr Adamowicz, klub Koalicji Obywatelskiej. Wysoka Izbo! Pytanie jest następujące: Czy należy nam przypominać, że Warszawa i Kancelaria Prezydenta leżą na śródlądziu? O tym wszyscy wiemy. Projekt tej ustawy szybko przesłałem do ludzi, którzy zajmują się przewozami morskimi. No niestety, w ich zgodnej opinii ten projekt wyklucza takie podmioty, jak Żegluga Gdańska, żegluga kołobrzeska, Żegluga Mazurska, żegluga szczecińska, operator obsługujący Kanał Elbląski. Te wszystkie podmioty są firmami polskimi.

Proszę, teraz pani poseł Mirosława Nykiel, klub Koalicji Obywatelskiej. Wysoka Izbo! To, że propozycja skalkulowana jest na kampanię Andrzeja Dudy, już padło wielokrotnie, i że dzieli, a nie łączy - to też. Ale do konkretów.

Zapewniono mnie 15 kwietnia, że prace trwają, że odbywają się spotkania i że będzie propozycja. 3 miesiące minęły i wyszły z tego nici, bo bon, który proponujecie, w żaden sposób nie rozwiązuje tego problemu. Moje pytanie brzmi: Gdzie są te nieprzebrane ilości gotówki, o której mówił Glapiński? Gdzie jest ta cudowna sytuacja budżetowa, o której mówił Morawiecki? I gdzie są [[Dzwonek]] te realne rozwiązania dla branży turystycznej? Proszę o zabranie głosu i zadanie pytania pana posła Piotra Borysa. Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! To blisko 4% PKB. 28 mld pozostawiają Polacy, blisko 45 mld - turyści z zagranicy. Żeby ratować polską turystykę, nie możemy jej dzielić. Dlatego już dzisiaj apelujemy do wszystkich państwa na tej sali sejmowej, także do Senatu, aby uwzględnić wszystkich Polaków: studentów, osoby pracujące, które mają dzieci powyżej 18. roku życia, osoby samotne, rolników i emerytów. Dlatego ta ustawa, jeżeli ma uratować z jednej strony branżę turystyczną, a z drugiej strony pozwolić na równość traktowania wszystkich Polaków, musi być dostępna dla wszystkich.

To jest po prostu niewybaczalne, dlatego będziemy apelować o uzupełnienie tej ustawy. Dziękuję bardzo panu posłowi. Wysoka Izbo!

Załogi są wysyłane na kwarantannę. Zaraz będą wracać całe załogi, całe jachty ze Szwecji od 13 czerwca przekonane, że jest otwarcie granic i jest zniesiona kwarantanna.

Macie dziury w systemie. Bardzo dziękuję. Pytanie zada pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pani minister.

Natomiast chciałabym spytać, jakie środki trafiły już do przedsiębiorców.

Dziękuję bardzo. Jeżeli na sali jest pan poseł Ireneusz Raś, a jest, prosimy, aby zabrał głos w celu sformułowania swojego wniosku. Dziękuję, panie marszałku.

Bardzo dziękuję panu posłowi. Niebawem odbędzie się Konwent Seniorów, gdzie w tej kwestii będzie podjęta decyzja.

To są rekordowe wzrosty, jakie notuje ta branża za naszych rządów, panie pośle. Moje pytanie, moje wątpliwości budzi to, skoro tak szeroko i aktywnie pan poseł dziś prezentuje tutaj swoje plany, jaką aktywnością pan poseł wykazywał się w czasie, kiedy Platforma Obywatelska kształtowała polityki publiczne.

Skoncentruję się przede wszystkim na tym elemencie i na tym wątku. Podczas prezentowania tutaj czwartej odsłony tarczy panowie i panie posłowie zarzucali nam, dlaczego poprawiamy kolejną ustawę, dlaczego nie zrobiliśmy jednej, doskonałej. Właśnie dlatego, żeby od 1 kwietnia pomoc trafiała na rynek natychmiast.

Odsunęliśmy o 180 dni możliwość. Mówię do pana posła, który zwrócił uwagę, że dopiero dziś. Nie, w pierwszej tarczy mieliśmy odsunięcie o 180 dni terminu koniecznego zwrotu za wydarzenia, które się nie odbędą. Oczywiście jest to rozwiązanie czasowe i nie jest ono ostatnim rozwiązaniem, jakie mamy dla branży turystycznej, z którą w ciągu ostatnich 3 tygodni spotykamy się regularnie co 2, 3 dni. Dla nich szyjemy kolejne rozwiązania, o nich też powiem za chwileczkę. Po pierwsze, w pierwszej tarczy już mieliśmy rozwiązania.

Z tarczy finansowej do branży turystycznej spłynęło już 4 mld zł. Czy państwo, panowie posłowie, wiedzą, jakie środki publiczne z samorządów, ze wspomnianego przez pana posła Miszalskiego Krakowa. Jak wygląda tarcza krakowska wsparcia turystyki, jak wygląda tarcza warszawska czy tarcza gdańska? Ona dzisiaj jest równa zeru. Te miasta nic nie zaproponowały. Skandal! ...w przeciwieństwie do Pragi, w przeciwieństwie do Wilna, w przeciwieństwie do portugalskiej Lizbony. Tam nic nie ma.

Jeszcze nie.

Beneficjentami tarczy będą wszystkie podmioty prowadzące działalność w ramach obszaru turystyka.

Każda jedna usługa turystyczna, która będzie finansowana, jest zapisana w tej ustawie. Zapraszam do skorzystania z ustawy, zapraszam do przeczytania.

Zatem beneficjentami będą np. organizatorzy - bo o tych też państwo pytali - wydarzeń kulturalnych, wydarzeń artystycznych, jeśli będą one częścią pakietu, także restauratorzy, nie wprost, nie bezpośrednio, ale nie jest to rozwiązanie przypadkowe. Przeanalizowaliśmy podobne rozwiązania obecne na Węgrzech, w Bułgarii, we Francji (Dzwonek) i we Włoszech.

Wątpliwości chciałabym przekazać.

Tak, proszę państwa, wiemy, co jest problemem branży turystycznej. Wiemy, że ona od pierwszego dnia kwarantanny, od 11 marca. najbardziej ucierpiała, ponieważ wtedy zaczęły się pierwsze anulacje wydarzeń turystycznych. Jednocześnie, jak powiedziałam, jest ona bardzo różnorodną branżą: od pojedynczych działalności gospodarczych, pilotów, przewodników, poprzez touroperatorów, wycieczki zagraniczne, hotelarzy i agroturystykę oraz kempingi.

Zatem ten bon będzie wspierał gospodarkę i będzie realnie pracował w gospodarce. Podział zaproponowany przez pana prezydenta dotyczy rodzin, to oznacza, że ponad 59% tej pomocy trafia do najuboższej części polskiego społeczeństwa. Trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś z państwa powiedziałby, że ta pomoc ma być w inny sposób dystrybuowana.

Proszę o zabranie głosu podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej panią minister Annę Surówkę-Pasek. Panie Marszałku! W pierwszej kolejności należałoby się odnieść do tego magicznego projektu o czeku turystycznym. Co z niego wynika? W zasadzie nic. Nie wiadomo, na jakich zasadach będzie przyznawany. Owszem, jest podany krąg beneficjentów, ale jest wskazana jakaś mitologiczna aplikacja, która będzie do tego służyła. Niestety wszelkie szczegóły dotyczące tego. kto będzie mógł go uzyskać, na jakich zasadach, jak będzie przebiegała rejestracja, kto będzie za to odpowiadał - to wszystko zostało odesłane do regulacji w drodze rozporządzenia. Problem polega na tym, że ta delegacja do uregulowania różnych absolutnie rzeczy w rozporządzeniu ma charakter czysto blankietowy, a jakkolwiek by na to popatrzeć, art. 92 polskiej konstytucji wyraźnie wskazuje, jakie elementy powinny być. Mało tego, polska konstytucja, na którą państwo się tak często powołujecie, wyraźnie wskazuje: to, co dotyczy dochodów, ma być uregulowane w ustawie, a tego tam nie ma. Co do wypowiedzi pana Kosiniaka-Kamysza powiem tak: brak różnicowania rzeczywiście miał miejsce. Wyrównanie wieku emerytalnego do 67 lat - rzeczywiście strzał w dziesiątkę, kompletny brak różnicowania. Natomiast odpowiadając na wszelkie pytania dotyczące wsparcia dla branży turystycznej: będzie to wsparcie dla polskich firm i tych, które w Polsce działają.

Proszę bardzo. I to, co słusznie tutaj wskazała pani premier: nie ma znaczenia ich formuła organizacyjna. Będą to również firmy, które świadczą te usługi w formie organizacji pożytku publicznego - stąd również PTTK będzie mogło z tego korzystać - a także firmy, które będą organizowały różnego rodzaju wydarzenia.

Warto o tym pamiętać. Co do samej wartości bonu - z projektu koalicji kompletnie nie wynika, czy będzie on zwolniony od podatku, czy będzie wliczany do dochodu, od którego zależy uprawnienie do nabycia innych świadczeń. Z projektu pana prezydenta wyraźnie wynika: jest on wolny od podatku, o czym stanowi art. 40 tego projektu, wolny od egzekucji komorniczej, niewliczany do wysokości dochodu, która będzie brana pod uwagę przy przyznawaniu różnego rodzaju świadczeń - art. 45. Natomiast pan prezydent konsekwentnie realizuje swoją politykę wsparcia dla Polaków, dla polskich rodzin. Doskonałym tego przykładem jest chociażby podpisanie ustaw, które wprowadzały trzynastą emeryturę, program 500+, który przecież wszedł w życie w 2016 r. Osoby, które osiągają dochód w tej wysokości, nie płacą w ogóle podatku. Natomiast warto również zauważyć, że podobne rozwiązania istnieją w innych państwach i są doskonałym wsparciem dla lokalnej branży turystycznej. Również bardzo ważne jest, że to jest projekt, który ma wesprzeć i polskie rodziny w zorganizowaniu wypoczynku, i przedsiębiorców, którzy w Polsce świadczą usługi turystyczne. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Pani Minister! Chcę powiedzieć, że bezpośredniego wsparcia branży turystycznej nigdy w Polsce nie było.

Bo pani o nim mówiła przez miesiące, ale pani go nie przygotowała.

Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o skierowanie projektu ustawy dodatkowo do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy za chwilę.

Wznawiam obrady. Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjęłam decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktu 3. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw, druki nr 203 i 405.

W takim razie bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku, żebyśmy sprawdzili, czy mamy kworum. Bardzo proszę.

Stwierdzam kworum. Powracamy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. W dyskusji zgłoszono wniosek o skierowanie projektu ustawy dodatkowo do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu jest, aby Sejm skierował ten projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu przyjął, a wniosek o dodatkowe skierowanie tego projektu ustawy poddam pod głosowanie. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za dodatkowym skierowaniem projektu ustawy zawartego w druku nr 423 do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym i senackim projektach ustaw o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druki nr 418, 283 i 419) Proszę panią poseł Urszulę Rusecką o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Przypadło mi w udziale przedstawienie sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny - sprawozdanie to druk nr 419 - o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, druk nr 418, oraz o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, druk nr 283. Wysoka Izbo!

Wielokrotnie byliśmy świadkami, jak Platforma Obywatelska, szczególnie w okresie wyborczym, składała Polakom obietnice bez pokrycia. I tak też było z tą złożoną w 2011 r. obietnicą o niepodwyższaniu wieku emerytalnego, złamaną tuż po wyborach. Bardzo proszę o przeniesienie dyskusji poza salę sejmową, aby pani poseł mogła przedstawić projekt. Proszę bardzo.

I to nie tylko złamane obietnice, ale także, jak myślę, zaplanowane oszczędności właśnie na emerytach. Przypomnijmy, że zlikwidowano emerytury pomostowe, podwyższono wiek emerytalny, chciano, by Polacy pracowali aż do śmierci.

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 16 czerwca 2020 r. projekt ustawy z druku nr 418 do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania.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 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tych projektów ustaw po posiedzeniu w dniu wczorajszym wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt ustawy. Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. I w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pani poseł Teresa Wargocka. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec projektów ustaw o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, senackiego zawartego w druku nr 283 oraz rządowego zawartego w druku nr 418, oraz sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zawartego w druku nr 419.

W ocenie trybunału zasada zaufania obywateli do państwa i prawa stanowionego nie może stwarzać pułapek dla obywateli. Ustawa obowiązująca od 2013 r. spowodowała, że kobiety, które przeszły na wcześniejsze emerytury, podjęły tę decyzję, nie mając świadomości, iż od tego momentu te emerytury są finansowane z ich składek i w ten sposób pomniejszają swój kapitał emerytalny. W momencie przejścia na emeryturę powszechną te emerytury otrzymały niższe, znacznie niższe. Ta niezgodność z konstytucją, przede wszystkim właśnie ta podstawa zaufania obywateli do państwa, do stanowionego przez państwo prawa, jest tymi projektami usuwana. Szanowni Państwo! To jest rozwiązanie, które spowoduje, że emerytury będą ponownie przeliczone i będą wypłacone różnice, czyli będzie wyrównana ta strata, która miała miejsce na przestrzeni tych lat. Mieliśmy dosyć długą dyskusję nad tymi projektami.

Można było nie oszczędzać na emerytach, nie sięgać do ich kieszeni. Można było zupełnie inaczej radzić sobie z kryzysem gospodarczym. Widzicie państwo teraz, jak rząd podchodzi do kryzysu.

Mówiła już pani przewodnicząca Rusecka o wieku emerytalnym. Kobiety, mężczyźni - 67 lat. 3 mln podpisów „Solidarności” do kosza. My to zmieniliśmy. Nie zrujnowaliśmy budżetu. Powrócił dawny wiek emerytalny. Skok na OFE. Kolejne 150 mld przepisane na konta ZUS-u. Nawet trybunał wam to klepnął, chociaż zabraliście pieniądze, choć obywatele uważali, że mają je na własnych kontach jako swoją własność. Przywróciliśmy to, zmieniliśmy to, zlikwidowaliśmy OFE.

Zaoszczędziliście na tych kobietach. Dzisiaj państwo mówicie, że to jakaś pomyłka, niedopatrzenie, wpadka. Ten wyrok wydał Trybunał Konstytucyjny w 2019 r., o którym wy, opozycja, mówicie: trybunał dublerów. Ten trybunał stoi na straży konstytucji i nawet ciężkie dla budżetu decyzje podejmuje zgodnie z duchem konstytucji.

Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska przedstawi pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz. Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Gdy pracuje się nad ważnymi zmianami, szczególnie w systemie emerytalnym, zdarza się, że można popełnić błędy. Ale najważniejsze jest, żeby umieć się do błędów przyznać. Jeszcze ważniejsze jest, żeby umieć je naprawić.

I teraz przechodzimy do orzeczenia, do wyroku, który wydał Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny nakazał tak naprawdę naprawić krzywdę wyrządzoną kobietom, szczególnie tym z rocznika 1953, które po prostu nie uzyskały w odpowiednim czasie informacji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących ich wysokości świadczenia i złożenia wniosków o emeryturę. Natomiast my, mając świadomość tego, że popełniliśmy błąd, chcieliśmy go jak najszybciej naprawić.

A, jeszcze jedno.

Bo wtedy nie było kampanii wyborczej. Szanowni Państwo!

W 2017 r. taka sama petycja w Senacie, również odrzucona głosami Prawa i Sprawiedliwości. W 2019 r. senatorowie przyjęli odpowiedni projekt, nawet bez zastrzeżeń waszego rządu, i ten projekt trafił nawet do Sejmu we wrześniu 2019 r., i nawet był w porządku obrad. Nie poddaliśmy się. I co się dzieje, szanowni państwo, kiedy on wpłynął? Otóż dalej, do dzisiaj właściwie go nie było. Pan marszałek, pan senator Marek Borowski trzykrotnie monitował u pani marszałek Wysokiego Sejmu, pani marszałek Witek, żeby ten projekt łaskawie dopuścić pod obrady. Ale tak się nie stało. I czego trzeba było, żeby ten projekt był w końcu tak naprawdę procedowany? Ano trzeba było kampanii wyborczej. Ano trzeba było spadających słupków poparcia dla urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Ale myślę, że nie o tym chcą słuchać emerytki, które czekają na ten projekt. My oczywiście jako Koalicja Obywatelska zagłosujemy za tym projektem. Nie widzimy powodu, dla którego tak naprawdę ponowne przeliczanie tych emerytur z urzędu ma następować dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Uważamy, że ten okres należy skrócić przynajmniej do 3 miesięcy.

Mało tego, one będą miały rację. Jeśli tu i teraz naprawimy ten błąd [[Dzwonek]] i poszerzymy ten krąg osób, to koszty dzisiaj będą dużo mniejsze niż te, które będą poniesione za jakiś czas. Dziękuję bardzo pani poseł, która zaprezentowała stanowisko klubu Koalicja Obywatelska. Proszę teraz o zabranie głosu panią poseł Karolinę Pawliczak, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czytając ten projekt ustawy, chce się powiedzieć: nareszcie. Nareszcie, po wielu miesiącach, a w sumie latach walki organizacji, ruchów społecznych, związków zawodowych, a przede wszystkim samych pokrzywdzonych przez tę wadliwą nowelizację ustawy z 2013 r., powoli sytuacja zmierza do właściwego jej uregulowania. Potrzeba uchwalenia projektowanej ustawy wynika nie tylko z konieczności wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale przede wszystkim z ułomności obowiązujących regulacji dotyczących postępowania o świadczenie emerytalno-rentowe. Z jednej strony to bardzo niepokojące, że dopiero ponad rok od wyroku trybunału sprawa ta doczekała się realizacji.

A błędy, jak pokazuje życie, mogą być popełnione, bo projekt ten niestety nie obejmuje wszystkich w imię zasady sprawiedliwości społecznej. Wszak w ocenie Trybunału Konstytucyjnego naruszona została zasada zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Oznacza ona konieczność w każdym, powtarzamy, w każdym przypadku zapewnienia bezpieczeństwa prawnego jednostki, a prawo nie może być pułapką na obywatela. Po to aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, że nie naraża się na skutki prawne, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania tych decyzji. Takiej możliwości została pozbawiona grupa osób urodzonych w 1953 r., które powszechny wiek emerytalny osiągały w okresie od lutego 2013 r. do kwietnia 2014 r., a więc w czasie, gdy obowiązywał już art. 25 ust. 1d. Ponadto uważamy, że słuszniejsze byłoby określenie zakresu podmiotowego ustawy bez ograniczenia wynikającego z odwołania się do rocznika 1953, odwołanie się bowiem do Trybunału Konstytucyjnego i do zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa można również odnieść do ubezpieczonych z innych roczników, którzy decydowali się na wcześniejszą emeryturę, ufając, że państwo nie zmieni reguł wypłaty powszechnego świadczenia emerytalnego. Dlatego przekazuję pani marszałek poprawkę klubu Lewicy dotyczącą zastosowania mechanizmu wzruszenia prawomocnych decyzji dotyczących zmiany art. 114 ustawy. Umożliwia ona uchylenie lub zmianę decyzji z powodu wadliwości bez ograniczenia czasu, jeśli w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji osoba zainteresowana nabędzie prawo do świadczenia lub świadczenie w wyższej wysokości. Pragniemy bowiem zapobiec w przyszłości takim problemom, z jakim mierzyły się osoby urodzone w 1953 r. Lewica mimo przekonania, że ten tryb jest niewłaściwy, będzie głosować za niniejszym projektem, bo uważamy, że grupa emerytów i rencistów i tak jest najbardziej poszkodowaną i ubogą grupą społeczną, którą należy wspierać. Nie godzimy się na jakiekolwiek nierówności w tej sprawie, bo chcemy sprawiedliwości, a grup wykluczonych, którymi należy zająć się natychmiast, jest przecież dużo więcej: to osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, którzy otrzymują jałmużnę, a nie wsparcie, wymieniać pewnie można byłoby dalej, bo nie należy już dłużej czekać. Wnioskujemy przy tym, aby po wejściu w życie tej ustawy tryb przyznawania świadczeń nie był znów złożoną i skomplikowaną procedurą. Prosimy o uproszczenie zasad oraz decyzji w stosunku do tych i tak już pokrzywdzonych osób. Dziękuję bardzo, pani poseł. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 przedstawi pani poseł Agnieszka Ścigaj. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W wyjaśnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest takie uzasadnienie. Trybunał Konstytucyjny powołuje się na zasadę zaufania do państwa, podkreśla, że prawo nie może być pułapką, przywilej nie może być pułapką.

To uzasadnienie skłania do głębszej refleksji i myślę, że ta refleksja powinna odnosić się do całego systemu emerytalnego.

Przecież takich sytuacji mamy wiele, bo jeżeli cały system opiera się na zastępowalności i ci, którzy wchodzą teraz w ten system, wiedzą, że za te 20, 30 lat tej zastępowalności po prostu nie będzie, to czy mogą mieć zaufanie do państwa i do tego systemu? Absolutnie nie, bo jak tutaj siedzimy, a przynajmniej moje pokolenie nie jest pewne, tak jak nie było pewne i otwartych funduszy emerytalnych, i zmian dotyczących różnych wcześniejszych możliwości, i tego, że na nasze emerytury. Czy nie jest to refleksja, która powinna być szerszą refleksją, tematem ponadpartyjnych rozmów na temat zmiany systemu emerytalnego, który absolutnie jest niewydolny? Czy nie taką pułapką było coś, co jest do tej pory nienaprawione, jak np. to, że matki, które opiekują się dzieciakami niepełnosprawnymi, matki na tzw. EWK, odeszły na emerytury, a po jakimś czasie pojawiła się możliwość innego świadczenia, i matki, które opiekują się dzieciakami, a nastąpiło to później, mają inne świadczenia pielęgnacyjne, mają wyższe kwoty, a ich emerytury dalej są niższe?

O to apeluję, i o to apeluje w tej chwili Koalicja Polska, żeby rzeczywiście ponadpartyjnie, ponadkampanijnie pochylić się nad systemem emerytalnym, bo on jest absolutnie niewydolny i nie daje poczucia bezpieczeństwa pokoleniom, a już szczególnie tym, którzy obecnie wchodzą w ten wadliwy system. 5 lat mija, prawie 6 lat - od niezrealizowanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który odnosi się do opiekunów osób niepełnosprawnych.

Być może to jest zbyt mała grupa wyborców i tę grupę można pominąć. Trzeba się nad tym pochylić. Proszę powiedzieć, czy te zasady, które są zawarte w tej ustawie, będą opierały się na uwzględnieniu zwaloryzowanych kwot składek emerytalnych, kapitału początkowego oraz wskaźnika długości życia adekwatnego do obecnego wieku osób uprawnionych do świadczeń.

Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła Michała Urbaniaka, który przedstawi stanowisko Koła Poselskiego Konfederacja. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Konfederacji.

Już za chwilę system, na którym się opieramy, ten system repartycyjny, będzie kompletnie niewydolnym systemem emerytalnym.

Słuszne jest to, by sprzątać bałagan - tutaj zwracam się do dobrej zmiany - ale, szanowni państwo, to dalej będzie tylko i wyłącznie łatanie dziury w tym już bardzo dziurawym suknie, z którego za chwilę po prostu może nic nie zostać. Potrzeba nam zmiany systemu opartego właśnie na wysokich składkach.

Dzięki temu coś, co dzisiaj nazywamy systemem trzeciofilarowym, będzie po prostu podstawą utrzymania się każdego Polaka na emeryturze. Kiedy mówimy też o systemie emerytalnym, powinniśmy pamiętać o demografii. To jest wręcz nierozłączne, te dwa obszary idą zawsze w parze. Czy rząd tak naprawdę planuje w ogóle jakiś kompleksowy program prodemograficzny? Wiemy, że to trudne. Żłobki, przedszkola, ulgi prorodzinne - to jest kierunek, w którym też powinniście iść. Bardzo dziękuję panu posłowi. Jeżeli nie ma więcej chętnych, to zamykam listę.

Wysoka Izbo!

Mówię tu o rządzie, a nie o Senacie oczywiście, który chce pewne rzeczy skutecznie naprawić. Pytanie zada teraz pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub parlamentarny Lewica. Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Kiedy wczoraj Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła ten projekt ustawy, wiele pań do nas napisało, uznając. Zacytuję te opinie: zasadne wydaje się zagwarantowanie jednolitych zasad zwrotu świadczeń należnych uprawnionym. Na taką potrzebę zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny.

Prosiłbym uprzejmie pana ministra, aby w swoim wystąpieniu jako osoba, która również reprezentowała Sejm, z tego, co wiem, przed Trybunałem Konstytucyjnym i która dzisiaj odpowiada (Dzwonek) za te kwestie, w sposób jednoznaczny wyjaśnił, czy przyjęty przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny projekt realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wprost, czy nadal pojawiają się te wątpliwości, o których mówiłem. Dziękuję. Pytanie zada teraz pani poseł Ewa Kołodziej, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Po pierwsze, gdzie państwo byliście, gdy w grudniu zeszłego roku do Sejmu trafił senacki projekt ustawy dotyczący emerytur kobiet z rocznika 1953? Gdzie państwo byliście, gdy pani marszałek podejmowała decyzję, by ten senacki projekt włożyć do zamrażarki?

Czy nie jest to może podyktowane względami politycznymi i wyborczymi?

W szczególności nie wiemy, czy wszystkie panie z rocznika 1953 będą potraktowane w jednolity, sprawiedliwy sposób i czy będą miały [[Dzwonek]] zagwarantowane jednolite zasady przeliczania i zwrotu zaległych świadczeń. Czy będą przygotowane odpowiednie regulacje, by tak właśnie się stało? Dziękuję bardzo. Pytanie zada teraz pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Nie widzę. Zatem teraz proszę pana posła Mieczysława Kasprzaka, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dzisiaj mamy dramat, jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne, o wysokość emerytur.

To jest bardzo niebezpieczne. Jest projekt obywatelski? Chodzi o zwolnienie pracujących emerytów z podatku. To jest ważne, to jest istotne, ale pytanie moje zmierza w kierunku.

Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Nie widzę na sali pana posła Mirosława Suchonia, zatem proszę o zadanie pytania panią poseł Małgorzatę Pępek, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sprawa ponownego przeliczenia wysokości emerytur dla osób z rocznika 1953 powinna być załatwiona już dawno temu. Dopiero kiedy pojawiła się kampania wyborcza, dopiero kiedy sondaże stały się dla Andrzeja Dudy niekorzystne, nagle przypomnieliście sobie o tej ustawie, po ponad roku od wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Według Najwyższej Izby Kontroli w zeszłym roku wydaliście na nagrody i premie prawie 400 mln zł.

Oczekują zdecydowanie więcej. Dlaczego kazaliście im czekać ponad rok? Skoro tak wam zależy na Polakach, to dlaczego nie skorzystaliście z senackiej ustawy, [[Dzwonek]] która wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego? Bardzo dziękuję. Pytanie teraz zada pani poseł Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Właściwie mam jedno krótkie pytanie.

Tutaj pojawiały się spory dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Ja mam wrażenie, że to jest zupełnie normalne, że w demokratycznych państwach Trybunał Konstytucyjny zajmuje się poprawianiem błędów legislacyjnych.

Dlaczego byliście państwo tak długo głusi na sprawy tych kobiet? Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zadanie pytania panią poseł Joannę Fabisiak, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Ułomność regulacji prawnych spowodowała krzywdę blisko 80 tys. kobiet. Bardzo dobrze, że próbujemy naprawić tę krzywdę. Ale czy naprawdę? Bo tam, gdzie jest istota tej ustawy, jest więcej niejasności niż faktów. Rzecz pierwsza, poruszana przez wiele osób. W uzasadnieniu czytamy, że tylko blisko 60 tys. kobiet skorzysta, mówiąc kolokwialnie, na tych zmianach ustawowych. Dlaczego te ponad 40% nie skorzysta? Znów jest niepokój. Jest jeszcze poważniejsza sprawa. Otóż słyszeliśmy, że wypłacana będzie różnica. Tak, ale jak będzie liczona ta różnica?

Bardzo proszę, panie ministrze, żeby pan nam przybliżył te fakty i żeby pan z tej trybuny uspokoił te kobiety, które przez tyle lat żyły z poczuciem krzywdy. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana posła Andrzeja Gawrona, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Czy to kampania, czy nie kampania, takie dobre ustawy trzeba przyjmować. W ostatnich miesiącach miałem wiele spotkań z osobami, które przychodziły do biura poselskiego i właśnie o tej sprawie mówiły, że trzeba to rozwiązać.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie teraz zada pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pierwsze pytanie podstawowe: Dlaczego tak długo trzeba było czekać, dlaczego trzeba było czekać na realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2019 r. To była podstawa do wznowienia postepowań, do zmiany decyzji ZUS-owskich. Te kobiety, dzisiaj 66-letnie, mają emerytury niższe nawet o 30% od kobiet o rok starszych lub młodszych, które pracowały tyle samo na podobnych stanowiskach.

Naprawdę to jest niegodne. Dzisiaj naprawiamy tę krzywdę. Dziękuję bardzo. Proszę zatem teraz pana Stanisława Szweda, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o odpowiedzi na pytania. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dotykamy bardzo trudnej i wrażliwej materii, jakim jest system emerytalny. Myślę, że wiele pytań, które padały tutaj, wynikało też z niezrozumienia tego systemu, który w Polsce funkcjonuje.

W tym zakresie Trybunał Konstytucyjny uznał, że jest to niezgodne z konstytucją.

Każdy oczywiście w innym zakresie, bo były różne momenty odchodzenia na emeryturę. Oczywiście ci, którzy przeszli na tę wcześniejszą emeryturę na starych zasadach, mieli wyższe emerytury, bo musimy powiedzieć, że funkcjonowali na zasadach starego systemu.

I teraz jeśli chodzi o te osoby, które nie złożyły. Mamy jedną zasadę w systemie ubezpieczeń: emerytura jest na wniosek pracownika. To nie jest przymus, to jest jego wybór.

Teraz dlatego jest ta różnica.

Oczywiście system emerytalny jest bardzo skomplikowany, on też - to, co mówiłem już w komisji - może spowodować, że ktoś, kolejna grupa, wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego z zarzutem, że jego stan jest gorszy od innych.

Ja mam dzisiaj wyliczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po posiedzeniu komisji jeszcze próbowaliśmy to jakoś wyliczyć.

Dlatego tak istotne i ważne są kwestie, które podejmujemy w systemie emerytalnym.

Bardzo dziękuję panu ministrowi. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 415 i 417) Proszę pana posła Kazimierza Smolińskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, druk nr 415.

Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu na posiedzeniu w dniu 17 czerwca br. wnosi, aby wysoki Sejm uchwalić raczył przyjęty projekt ustawy. W trakcie dyskusji na posiedzeniu komisji zgłoszono, jeden z klubów zgłosił projekt zmiany w tym projekcie. Chodziło m.in. o to, aby odtajnić wszelkiego rodzaju akta czy teczki, jak to się mówi, trzymane w Instytucie Pamięci Narodowej. W związku z tym, że zgodnie z opinią prawników sejmowych, zresztą jest tak też w przekonaniu większości członków komisji, wykracza to poza zakres rozstrzygnięcia, które jest przedmiotem dzisiejszej debaty czy dzisiejszego czytania, komisja negatywnie zaopiniowała te zmiany.

Natomiast dzisiejsze przedłożenie jest potrzebne, aby te zbrodnie komunistyczne, które nie są zbrodniami wojennymi, nie uległy przedawnieniu, ponieważ z dniem 1 sierpnia br. to przedawnienie by nastąpiło, natomiast jeżeli chodzi o te pozostałe zbrodnie komunistyczne, to przedawnienie nastąpiłoby za 10 lat.

Projekt został przyjęty w tym kształcie, który jest Wysokiej Izbie przedstawiony. Proszę, tak jak wnosiłem, o przyjęcie tego projektu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Proszę panią poseł Annę Milczanowską o przedstawienie stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Przedmiotem i istotą proponowanych przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości zmian w obowiązującym porządku prawnym jest przede wszystkim umożliwienie bezwzględnego i nieograniczonego czasem ścigania zbrodni komunistycznych, a tym samym niedopuszczenie do możliwości przedawnienia karalności tychże zbrodni, co zgodnie z obowiązującą ustawą nastąpiłoby 1 sierpnia tego roku. W świecie wartości, którym hołdujemy, pewność i nieuchronność kary za zbrodnie popełnione przeciwko człowiekowi nie stanowią przedmiotu sporu. U podstaw funkcjonowania demokratycznego państwa stoi pewność obywatela co do posiadania fundamentalnych praw, u których źródła leży ludzka godność. Dlatego ściganie oprawców komunistycznych, którzy sprzeniewierzyli się istocie człowieczeństwa, nie może być ograniczone jakąkolwiek datą. Powołany ustawą z grudnia 1998 r. Instytut Pamięci Narodowej od lat zajmuje się ściganiem nazistowskich i komunistycznych zbrodniarzy, przywraca cześć żołnierzom i bohaterom codziennej walki o Polskę. Podczas posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości, która niemal w całości zaaprobowała przedmiotowy projekt ustawy, reprezentujący Instytut Pamięci Narodowej prokurator Robert Kopydłowski przedstawił informację, że w Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prowadzonych jest obecnie 431 postępowań w sprawach o zbrodnie komunistyczne, a w ponad 300 zastosowano kwalifikację z art. 3 jako zbrodnie przeciwko ludzkości. Szanując pamięć komunistycznych zbrodni, musimy dzisiaj zrobić wszystko, by winni ponieśli odpowiedzialność za swoje czyny. Brak zgody na przedawnienie ścigania i sądzenia zbrodniarzy znajduje podstawę zarówno w polskiej konstytucji i mądrej polityce kryminalnej państwa. Dlatego Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość jest zdecydowanie za przyjęciem tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo, pani poseł. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska głos zabierze pan poseł Michał Szczerba. Szanowny Panie Marszałku!

Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć: oczekiwaliśmy w tej sprawie projektu rządowego, projektu, który powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości, projektu wyprzedzająco przygotowanego, który nie pozwoli na to, że od 1 sierpnia zbrodniarze komunistyczni nie będą w sposób należyty osądzeni. Wiemy, że to ministerstwo, Ministerstwo Sprawiedliwości, słynęło z różnych nowelizacji ustawy o IPN. One powodowały wyjątkowe wzburzenie w obszarze stosunków międzynarodowych, spowodowały różnego rodzaju konsekwencje, z których później rząd musiał wycofywać się rakiem. Szanowni Państwo! Kwestia, którą się zajmujemy, kwestia, którą klub Koalicji Obywatelskiej w pełni popiera, ma jeden podstawowy cel, aby te zbrodnie, aby te przestępstwa się nie przedawniły. Szanowni państwo, czym są zbrodnie komunistyczne?

Polegają one na stosowaniu represji lub innych form naruszenia praw człowieka wobec jednostki lub grupy ludności bądź w związku z ich stosowaniem. I one stanowią przestępstwo według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie jego popełnienia. Ale również są innego rodzaju przestępstwa, które nie były sankcjonowane przez państwo komunistyczne, a śledztwa, które prowadzi IPN, prowadzi komisja ścigania zbrodni, mogą zakończyć się sformułowaniem aktu oskarżenia. Również oczekiwaliśmy, i mówię to jako przedstawiciel Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, że instytucja, jaką jest IPN, której budżet wzrósł w sposób znaczący, tj. z 250 mln w 2015 r. do 350 mln w roku 2020, będzie nas jako władzę ustawodawczą informowała o tego typu niebezpieczeństwach, bo przecież w tej chwili tylko sprawne procedowanie i pełne wsparcie dla tej inicjatywy legislacyjnej może zagwarantować to, że zbrodniarze nie unikną należnej odpowiedzialności. Wydawało się, że IPN powinien o tej sprawie nas informować. Kolejna sprawa. Chcielibyśmy również, żeby akta komunistycznych służb były aktami jawnymi. Nie może być tak, że jacyś politycy, jacyś funkcjonariusze są wyłączeni z tych działań instytucji państwowej.

Nie ma również naszej zgody na to, żeby cały aparat państwa był zaangażowany w to, że komunistyczny prokurator, który był przez chwilę również posłem na tej sali, będzie udawał, że jako prokurator komunistyczny był ofiarą tego systemu, którego był funkcjonariuszem, ale również od którego otrzymywał odznaczenia państwowe. Nie może być również tak, żeby powtórzyło się kiedykolwiek, że prezes funduszu państwowego nagle nie odnajduje się na liście osób, które podlegają ustawie lustracyjnej, tylko i wyłącznie dlatego, że na początku lat 90. robił interesy (Dzwonek) z prezesem ważnej partii politycznej. Chciałbym bardzo jednoznacznie powiedzieć: zrobimy wszystko - i tu, jako opozycja parlamentarna, ale również jako większość prodemokratyczna w Senacie - aby te przepisy zaczęły obowiązywać 31 lipca i żeby od 1 sierpnia, tak jak do tej pory, komunistyczni zbrodniarze nie mogli czuć się bezpieczni. Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Maria Żukowska przedstawi stanowisko klubu parlamentarnego Lewica. Wysoka Izbo! Najpierw parę słów o instytucji, o której będziemy mówili, o Instytucie Pamięci Narodowej. Lewica od wielu lat, od początku mówi, dlaczego opowiadamy się za likwidacją IPN-u. Myślę, że najtrafniej uzasadnił to prof. Andrzej Romanowski, były naczelny „Polskiego słownika biograficznego”, również były działacz „Solidarności”: Instytut Pamięci Narodowej łączy pod jednym dachem dwie instytucje: prokuraturę i placówkę historyczną. A przecież cele obu instytucji są całkowicie odmienne. Prokurator zmierza do osądzenia, historyk - do zrozumienia mechanizmów. Prokurator nie szuka okoliczności łagodzących - nad tym może się zastanawiać adwokat, i to nie w IPN, bo tam go nie ma, lecz na rozprawie sądowej. Historyka natomiast nie interesuje kwestia winy czy kary, lecz analiza procesu dziejowego. IPN zniszczył życie wielu osobom. 50 tys. funkcjonariuszy straciło emerytury. Czy byli to zbrodniarze? W tej grupie są sprzątaczki w szpitalu MSW, kierowcy, twórcy bazy PESEL, SOK-iści, pogranicznicy. Będziemy walczyć o przywrócenie im godnych emerytur. Złożyliśmy już projekt ustawy w tej sprawie. Ale wracając do tematu IPN-u: Co zrobić z masą likwidacyjną po IPN-ie? Bo mamy taki zamiar, żeby oczywiście IPN przestał dalej funkcjonować. Archiwalia powinny zostać przekazane do Archiwum Akt Nowych. Edukacja historyczna powinna być realizowana w postaci grantów badawczych, o które ubiegają się uniwersytety i inne instytucje naukowe. Biuro Lustracyjne powinno zostać zlikwidowane - niech kwestie związane z agenturą badają historycy.

Dla porównania budżet Państwowej Akademii Nauk to 83 mln zł. Czyli w ostatnim roku IPN dostał od PiS podwyżkę, która przewyższa budżet całej Polskiej Akademii Nauk. Macie tyle pieniędzy, że sami nie wiecie, na co je wydawać. Na co idą te setki milionów złotych? Według NIK prokurator w IPN-ie zarabiał średnio 18 tys. zł miesięcznie w 2018 r. Lewica nie sprzeciwia się ściganiu przestępstw popełnionych w okresie PRL. Jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, powinien być osądzony przed sądem demokratycznej Polski. Takie jest stanowisko polskiej lewicy od 30 lat.

Dziś także chcę powiedzieć, choć być może nie ja powinienem to mówić, tym wszystkim, a oni są też na tej sali, którzy doświadczyli krzywd i niegodziwości władzy i systemu przed 1989 r.: przepraszamy. Te słowa nadal obowiązują. Odrzuciliśmy system, bronimy ludzi i wartości. Każdego dnia będziemy bronić ludzi przed odpowiedzialnością zbiorową, ale jeśli zbrodnie zostały popełnione - nieważne, czy w latach 50., czy 80. - to winni muszą zostać ukarani. Dlatego klub Lewicy złoży swój projekt ustawy o IPN-ie, natomiast poprze przedłożony przez Prawo i Sprawiedliwość projekt ustawy. Dziękuję bardzo. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 przedstawi pan poseł Jacek Protasiewicz. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Koalicji Polskiej jest jednoznacznie za tym, ażeby zbrodnie komunistyczne nie ulegały przedawnieniu. Dlatego uważamy ten projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za projekt jak najbardziej zasadny, zwłaszcza że rzeczywiście z końcem następnego miesiąca, 31 lipca tego roku, przedawnieniu uległyby te zbrodnie komunistyczne, które nie są zbrodniami zabójstwa, ale - jak to zostało już wyjaśnione w jednym z wcześniejszym wystąpień - oznaczały stosowanie represji i naruszanie praw człowieka w okresie istnienia PRL-u, a tych przypadków było wiele i nie wszyscy, którzy się tego dopuszczali, zostali właściwie osądzeni.

Piękne słowa, ale jak one mają się do rzeczywistości? Jak mają się do tego, że to w państwa szeregach, z państwa rekomendacji osoby uwikłane w system opresji z czasów państwa komunistycznego, osoby, w przypadku których udowodniono albo istnieją namacalne dowody, że brały udział w tym, co jest w ustawie o IPN zdefiniowane jako zbrodnia komunistyczna - chodzi o represje i naruszanie praw człowieka - nie tylko nie ulegają karze, ale są wynagradzane stanowiskami i prominentnymi pozycjami w systemie instytucjonalnym wolnego państwa Rzeczypospolitej Polskiej?

Jest przypadek sędziego Iwulskiego, którego aktualny prezydent Andrzej Duda w 2016 r. powołał na prezesa jednej z izb Sądu Najwyższego, a to jest sędzia, który w okresie stanu wojennego, czynny, w mundurze wojskowym, wydawał wyroki na działaczy opozycyjnych. Skazano z jego udziałem 16 osób, w tym 13 - na kary więzienia. Chwała Bogu, że już jej nie ma na tej sali. Przez lata był senatorem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, a w stanie wojennym - prokuratorem stanu wojennego.

A więc deklaracje - jedno, piękne słowa o wartościach - drugie, a rzeczywistość, niestety - bardzo przykra. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo!

Apelujemy również o to, żeby ujawnić aneks do raportu o WSI. Apelujemy o to. Apelujemy o to, żeby to się wreszcie dokonało, bo mija 5 lat kolejnej prezydentury i nie ma tego aneksu. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Natomiast jeśli chodzi o dekomunizację w Polsce, to niestety III RP nie przeprowadziła dekomunizacji, tę dekomunizację przeprowadza dopiero biologia. Dopiero biologia przeprowadza w Polsce dekomunizację. Co do Instytutu Pamięci Narodowej - niestety nie spełnia on do końca swoich zadań, o czym mówił wielokrotnie też Krzysztof Bosak jako kandydat na prezydenta, zwracając uwagę, że chociaż w zapisach ustawy o IPN jest wprost określone, że ma on bronić dobrego imienia Polski i Polaków, to np. nie ma regularnie prowadzących polemikę anglojęzycznych kont w mediach społecznościowych IPN-u, które by non stop prowadziły tego typu prace. To jest ogromne zaniedbanie.

O tym projekcie nie kto inny jak premier Beata Szydło mówiła: Nie ma w niej niczego, co godziłoby w nasze relacje czy poszukiwanie prawdy i mówienie o niej w tym rozumieniu, o którym mówi państwo Izrael. Podkreśliła, że Holokaust był wielką tragedią wywołaną przez Niemców i należy ścigać wszystkich, którzy to kwestionują. Ta ustawa wreszcie kończy z tym, że można bezkarnie kłamać na temat tego, że były polskie obozy śmierci. To nieprawda. To są słowa pani premier Beaty Szydło z marca 2018 r., po ustawie ze stycznia 2018 r.

Szczęść Boże! Szczęść Boże w ciężkiej pracy dla ojczyzny wszystkim pracowitym, prawdomównym, szukającym prawdy o naszej historii pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej! Nie lękajcie się. Tak długo, jak długo w Sejmie zasiadają posłowie koła Konfederacja, które oby urosło do rozmiaru klubu, nie lękajcie się pogróżek ze strony Lewicy, która wprawdzie koniunkturalnie głosować będzie za tym projektem, ale wygraża wam, wraz kolegami z innych klubów grozi likwidacją tej zasłużonej dla poszukiwania i kultywowania pamięci historycznej Polaków instytucji. Teraz ta ustawa, nad którą dzisiaj tutaj procedujemy. Jasna sprawa, bez przedawnienia w przypadku zbrodni komunistycznych, sowieckich, niezależnie od tego, czy w rosyjsko-, czy w polskojęzycznym wydaniu, czy też w jidysz, który był językiem popularnym w niektórych instytucjach zbrodni na narodzie polskim, bez różnicy. Zbrodnie komunistyczne bez przedawnienia.

I jeszcze jeden szczegół, panie marszałku, pani marszałek, przepraszam, nastąpiła zmiana. W dniach, w których fałszowanie historii przybiera wymiar instytucjonalny, głowy państw, w tym prezydent Federacji Rosyjskiej, nie wahają się przypisywać Polsce odpowiedzialności za rozpętanie II wojny światowej, jest szczególnie ważne, żebyśmy tutaj, w Warszawie, byli jednoznaczni w ocenie zbrodni komunistycznych i udziału Związku Sowieckiego w rozpętaniu II wojny światowej. Przechodzimy do pytań. Wyznaczam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Zamykam listę posłów chętnych do zadania pytania. Bardzo proszę. Szeregowy Pośle Kaczyński! W uzasadnieniu do tej ustawy wnioskodawcy powołują się na fragment preambuły konstytucji, podkreślają, że dbając o prawa człowieka, chcą bezterminowo ścigać zbrodnie komunistyczne. Nie mam nic przeciwko temu, ale pragnę zapytać: Kiedy zajmiemy się dzisiejszym łamaniem praw człowieka przez rządzących? Kiedy przestaniecie przymykać oko na to, że studenci Uniwersytetu Śląskiego od kilku tygodni są przesłuchiwani na policji, bo nie zgadzali się z katolicką ideologią na świeckiej uczelni i homofobicznymi wypowiedziami jednej z wykładowczyń? Kiedy przestaniecie wykorzystywać pandemię do tego, by zabraniać ludziom zgromadzeń, gdy są dla was niewygodne, podczas gdy wasz rząd mógł w szczycie zachorowań się spotykać, gdzie chciał, jak chciał i w jakim składzie chciał?

Proszę zająć się poważnymi sprawami, śledzić obrady Sejmu i zadawać. Pani poseł, przywołuję panią do porządku. Bardzo proszę. Aha, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Nie widzę. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Osądzenie zbrodni komunistycznych ma nie tylko wymiar prawny, lecz stanowi również wyraz potępienia moralnego dla takich czynów, ugruntowania w świadomości społecznej ich karalności, a także zapewnienia pokrzywdzonym, ich rodzinom i całemu społeczeństwu poczucia sprawiedliwości. Dopuszczenie do przedawnienia zbrodni komunistycznych stanowiłoby natomiast zaprzeczenie wartościom konstytucyjnym oraz powszechnie uznawanym przez społeczność międzynarodową. Mam pytanie do wnioskodawców, ewentualnie do przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości czy IPN-u. Otóż ten projekt ma dotyczyć jedynie postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 423 mln zł ma kosztować w bieżącym roku wszystkich podatników funkcjonowanie IPN-u. To o 63 mln zł więcej niż w roku minionym. Dla porównania Państwowa Inspekcja Pracy, która powinna stać na straży tego, aby ludzie w pracy czy ludzie pracy w Polsce byli zatrudnieni zgodnie z prawem i aby ich praca była bezpieczna, dostaną tylko 374 mln zł. Dr Jarosław Szarek, prezes IPN-u, w jednym z wywiadów stwierdził, że IPN bardzo dba o odpowiednią edukację młodzieży, aby w przyszłości mogła stanowić elitę naszego narodu. Działania przyjmują różną formę: od wystaw, audiobooków aż po gry i komiksy. Chciałem dowiedzieć się, ile milionów z publicznych środków zostało wydanych na różnego rodzaju gry planszowe. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Według Lewicy IPN należy zlikwidować, archiwalia, teczki przekazać do Archiwum Akt Nowych.

Nie grajmy teczkami. Dość grania teczkami, tak jak w przypadku byłego prezydenta Lecha Wałęsy - okazało się, że z dużej chmury mały deszcz. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Przypomnę dane już podane przez przedstawicielkę Lewicy. Budżet Państwowej Akademii Nauk - 83 mln, budżet IPN - 423 mln, liczba pracowników PAN - 8700, liczba pracowników IPN - 2200. IPN dostaje kilkadziesiąt milionów złotych więcej niż Państwowa Inspekcja Pracy.

Średnie wynagrodzenie naukowczyni czy naukowca w PAN to nieco ponad 3 tys. zł, średnie wynagrodzenie pracownika jest dokładnie dwa razy wyższe, to ponad 6 tys. zł. Śledztw mniej, zarobki coraz wyższe. Jakbyście płacili tyle Państwowej Akademii Nauk, to wszystkie zbrodnie byłyby już udokumentowane. Jakbyście płacili tyle samo prokuratorom, to wszyscy zbrodniarze siedzieliby już w więzieniach. Jaka jest wydajność? Jak liczymy opłacalność funkcjonowania takiej instytucji jak IPN? Czy nam się to po prostu [[Dzwonek]] opłaca: ściganie i dokumentowanie w wydaniu IPN? Pani poseł Monika Falej, klub Lewica. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Mam kilka krótkich pytań. Po pierwsze, czy kolejne 30 lat będą ukrywane teczki?

To są przestępstwa właśnie przeciw Polkom i Polaków i to jest bardzo ważne. Dziękuję. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mówimy dzisiaj o ustawie, która ma ścigać zbrodniarzy. I to dobrze, bo jako Lewica uważamy, że nie może być tak, że ktoś pozostaje bezkarny. 423 mln przeznaczyliśmy w tym roku na IPN.

Moi znajomi, przyjaciele z Jeleniej Góry, Legnicy, Bolesławca czy Zgorzelca zostali pozbawieni prawa. Do emerytury.

Bardzo proszę.

Wysoka Izbo!

Przecież macie państwo świadomość, jak wiele krzywdy z tego powodu się dzieje, jak wiele osób.

Człowiek, który jest niewinny, potem, po powtórnym badaniu otrzymuje informację, tak, nie był współpracownikiem, tak, jest niewinny itd. Jaki jest powód tego, że jest ta niepotrzebna tajemnica? Mówicie państwo często o tym, że prawda jest najważniejsza, a więc ujawnijmy tę prawdę (Dzwonek), pozwólmy każdemu stanąć w obliczu prawdy o sobie samym. Dziękuję bardzo, pani poseł.

Uważamy, że nie powinny ulegać przedawnieniu zbrodnie komunistyczne. Martwi mnie tylko, że tak ważny projekt, o którym Prawo i Sprawiedliwość mówi jako kluczowym dla siebie, procedowany jest właśnie w taki sposób: jako projekt poselski, w ostatniej chwili, niemalże z ryzykiem, że ta zmiana mogłaby nie wejść w życie. Zdecydujcie się, co jest naprawdę ważne, i przestańcie zajmować się sprawami, które są nieistotne, i skupcie się na rozwiązaniach, które wymagają tego, żeby były rozpatrywane we właściwym czasie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo cieszy mnie fakt, że taki projekt jest teraz w parlamencie. Trzeba pamiętać o tym, że wszelkie zbrodnie komunistyczne, jakie miały miejsce, to są rzeczy, o których nie wolno zapominać. Możemy przebaczać, ale nigdy nie zapominajmy o tym, co komuna zrobiła z narodem polskim. Cieszę się, że taki projekt będzie pozwalał na to, aby dalej ścigać zbrodniarzy komunistycznych, ale mam też bardzo konkretne pytanie. Gdzie ujawnienie raportu WSI przez prezydenta? Tego nie ma, a powinno być już dawno zrobione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Na postawione pytania odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pan minister Marcin Warchoł. Zapraszam, panie ministrze. Było jedno pytanie do nas. Odpowiadam panu posłowi Sonikowi.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. W imieniu posłów wnioskodawców na pytanie odpowie pani poseł Anita Czerwińska. Zapraszam, pani poseł. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Proszę państwa, z jednej strony cieszy jednomyślność, która była już na posiedzeniu komisji. Wszyscy państwo wypowiedzieli się w ten sposób, że popierają tę ustawę. No może z jednym wyjątkiem. Jako jedyny wstrzymał się poseł Konfederacji. Więc panowie, jak mówicie, że chcecie dekomunizacji, to bardzo proszę: czyny, nie słowa. Bo na tej mównicy można powiedzieć wszystko, ale my, poprzez głosowanie oświadczamy i deklarujemy, czego naprawdę chcemy i oczekujemy. Więc jeśli chcecie dekomunizacji, to zagłosujcie za tym. Proszę państwa, z jednej strony cieszy ta jednomyślność, ale z drugiej strony martwi, że niektórzy państwo posłowie nie rozumieją tej ustawy i nie rozumieją, jak jest skonstruowany Instytut Pamięci Narodowej. Pani poseł, wiem, że nie jest pani w tej komisji, nie była pani na posiedzeniu. Otóż Instytut Pamięci Narodowej to jest Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, to jest ten pion śledczy, który właśnie zawiera się w tej ustawie, a kwestie, które porusza pani czy też poruszaliście państwo, dotyczą innych pionów, wydziałów i biur Instytutu Pamięci Narodowej, czyli Archiwum, czyli Biura Lustracyjnego i Biura Edukacji Publicznej. Więc ja bardzo bym prosiła, żeby kwestii, które państwo podnoszą, jakby nie wkładać do tej ustawy, bo już na posiedzeniu Sejmu prawnicy odpowiedzieli państwu, że to wychodzi poza zakres przedłożenia. Więc dyskutujmy o tych sprawach, bo rzeczywiście dekomunizację trzeba w Polsce skutecznie przeprowadzić, ale bardzo proszę, żebyśmy [[Oklaski]] nie wprowadzali w błąd siebie nawzajem, no a przede wszystkim opinii publicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu przedstawienia sprawozdania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 421) Proszę panią poseł Barbarę Bartuś o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W polskim systemie władza prawa władza ustawodawcza należy do Sejmu i Senatu. Funkcja prawodawcza jest jedną z trzech podstawowych funkcji Sejmu. Polska konstytucja nie przewiduje możliwości zastępowania Sejmu w jego funkcji ustawodawczej przez inne organy. Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 marca br. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dodano do regulaminu Sejmu dział IIIa zawierający przepisy określające zasady odbywania posiedzeń Sejmu, komisji i podkomisji sejmowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

Parlamenty w całym regionie OBWE muszą zatem podjąć zdecydowane kroki, aby zapewnić kontynuację prac w okresie blokady i dystansu społecznego. Widzimy, że wiele z parlamentów właśnie to robi. Pomimo zakłóceń harmonogramów i trudności w organizowaniu regularnych sesji plenarnych i komisji, co wpływa na spowolnienie regularnego procesu stanowienia prawa, liczne parlamenty w całym regionie OBWE wykazują elastyczność i zaangażowanie w dostosowaniu się do bieżących okoliczności. Niektóre parlamenty podjęły szybkie działania w celu zmiany swoich regulaminów wewnętrznych lub sposobu uchwalania ustaw, które pozwalają im kontynuować działalność za pośrednictwem platform internetowych i pracy zdalnej. W innych krajach po raz pierwszy internetowe spotkania komisji parlamentarnych są transmitowane na żywo w Internecie i telewizji, dzięki czemu sytuacja nadzwyczajna staje się okazją do zwiększenia przejrzystości, zobrazowania odpowiedzialności oraz przybliżenia pracy parlamentarnej obywatelom w czasach, gdy wielu czuje się niedoinformowanych i odizolowanych. Ten komunikat wydany przez OBWE blisko miesiąc po tym, jak wprowadziliśmy te przepisy, można uznać za pochwałę polskiego Sejmu. Mało tego, ten komunikat był zobrazowany zdjęciem z polskiego Sejmu.

Dlatego też ten rozdział stosuje się tylko do takich sytuacji. Ten rozdział nie nakazuje trybu zdalnego, tak jak powiedziałam, poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej, tylko ten artykuł, te przepisy mówią, że w zaistnieniu jednej z tych sytuacji posiedzenie Sejmu może być prowadzone z wykorzystywaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

Taka jest nasza rekomendacja i wydaje się, że ten przepis może istnieć, [[Dzwonek]] a to, czy on będzie wykorzystywany, będzie zależało od sytuacji, jaka będzie panowała w naszym kraju. Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Kazimierz Smoliński. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec poselskiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, druk nr 421. Zmiana regulaminu, która jest proponowana, tak jak to przedstawiła pani poseł wnioskodawczyni, zmierza do uchylenia art. 2, który wprowadza czasową możliwość przeprowadzania zdalnych posiedzeń Sejmu i zdalnych posiedzeń komisji, które może zwoływać marszałek Sejmu. Naszym zdaniem jest to rozwiązanie słuszne. Przedstawiając to rozwiązanie kilka miesięcy temu, wychodziliśmy z założenia, że po kilku miesiącach skończy się czas pandemii. Niestety wbrew niektórym politykom rząd nie wie, kiedy stan pandemii się skończy.

Dziękuję bardzo. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi Wysokiej Izbie pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska. Bardzo proszę. Panie i Panowie Posłowie! Proszę mi powiedzieć, jak to jest: pielęgniarki mogą, lekarze mogą, kolejarze mogą, fryzjerzy mogą, górnicy mogą - wszyscy mogą. Odmrażamy gospodarkę, pracujemy, staramy się, zachowując pewne rygory sanitarne, funkcjonować normalnie, i nagle oto w Sejmie Rzeczypospolitej jest taka grupa, lepsza grupa, może to lepszy sort.

Dobrze, zdołaliśmy się do tego przyzwyczaić. Tylko chcę powiedzieć, że to nie jest ta zmiana w regulaminie o umożliwieniu zdalnego porozumiewania się za pomocą urządzeń elektronicznych. To jest o tym, że nie mamy inicjatywy zwoływania komisji, nie mamy inicjatywy zwoływania podkomisji, że wszystko jest w rękach pani marszałek. Nie ma dyskusji, nie ma ekspertyz, nie ma gości na posiedzeniu komisji. To się staje Sejm niemy.

Państwu Sejm nie jest do niczego potrzebny. Wy macie kłopoty. Połowa waszego klubu, mówię tu do Zjednoczonej Prawicy, to są członkowie rządu. To gdzie oni mają czas siedzieć tu, głosować, dyskutować? A tak, zdalnie, zawsze jest jakiś gabinet polityczny, sekretarka, ktoś to wykona, głosowania mają znakomitą frekwencję. Opozycja nie zabiera głosu, opozycja nie piętnuje, opozycja nie składa wniosków, opozycji nie ma. Państwo potraktowaliście Sejm jako gospodarstwo pomocnicze rządu. Państwu Sejm do niczego nie jest potrzebny. To niedługo nasze dzieci i wnuki będą miały w podręcznikach historii taką definicję: Sejm - zespół budynków w centrum Warszawy o ciekawej architekturze niedaleko kościoła pw. św. Aleksandra. Nie ma na to naszej zgody.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie Polaków klub Lewica od samego początku stanu zagrożenia epidemicznego i późniejszego stanu epidemii wspierał wszystkie działania rządu zmierzające do ograniczania skutków rozprzestrzeniania się COVID-19. Z tego też względu, w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie posłów i posłanek, a także w trosce o zapewnienie ciągłości funkcjonowania Sejmu, przychyliliśmy się do wniosku o wprowadzenie do działu III regulaminu Sejmu możliwości odbywania posiedzeń Sejmu, komisji i podkomisji sejmowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Wyrażenie zgody na taki tryb pracy Sejmu było z naszej strony gestem dobrej woli. Nie oznacza to jednak, że nie mieliśmy obaw przed podjęciem takiej decyzji. Mamy bowiem świadomość, że Prawo i Sprawiedliwość w praktyce bardzo ostrożnie gospodaruje prawem, a tym bardziej sprawiedliwością. Są jednak w życiu sytuacje nadzwyczajne, w których odpowiedzialne siły polityczne, rzeczywiście dbające o dobro obywateli i obywatelek wznoszą się ponad doraźne, partykularne interesy, słupki poparcia czy spokojny sen prezesa. Sądziliśmy, że w obliczu bezprzedmiotowego zagrożenia pandemią COVID-19 wyciągnięta przez nas w geście dobrej woli ręka spotka się z życzliwym i pełnym zrozumienia przyjęciem, a tymczasem ona nie raz została dotkliwie pogryziona, i tylko z niewielką satysfakcją trzeba przyznać, że nie została odgryziona. Możliwość odbywania posiedzeń Sejmu, komisji i podkomisji sejmowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej niejednokrotnie przekraczała granice dobrego parlamentarnego obyczaju. Posiedzenia komisji zwoływane są z dnia na dzień pod dyktando partii rządzącej, kalendarza wyborczego czy oczekiwań zwykłego posła. W takich warunkach nie da się zaplanować rzetelnej pracy w okręgach, nie da się uczciwie i odpowiedzialnie przygotować do obrad czy pracy w komisjach. Naprawdę nie wszyscy posłowie i posłanki mieszkają w stolicy czy, precyzyjnie mówiąc, na elitarnym Żoliborzu. Wiele zastrzeżeń mamy do prac w komisjach. Obserwujemy, że w komisjach podczas głosowań telefonicznie mobilizowani do oddania głosów są posłowie partii rządzącej i dopiero po oddaniu przez nich głosów procedura głosowania jest zakańczana. To nie jest dobra praktyka. Rząd i minister Szumowski systematycznie odmrażają kolejne sfery życia publicznego. Klienci wrócili do galerii handlowych, uczniowie napisali matury, wierni wrócili do kościołów, żałobnicy - na cmentarze, kibice - na trybuny, a 460 posłów i posłanek [[Dzwonek]] nie może wrócić do pracy, za którą dobrze wynagradzają ich podatnicy. Lewica stanowczo opowiada się za przywróceniem obrad Sejmu w trybie sprzed epidemii. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Jarosław Sachajko. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Przepraszam bardzo, panie pośle. Jeśli państwo chcecie się kłócić, to poza salą plenarną. Bardzo proszę. Przedstawiony druk w obecnym brzmieniu, w lakonicznym trzylinijkowym tekście ma zalegalizować dalsze bezterminowe zdalne i ograniczone w swojej formie prowadzenie prac Sejmu. Wysoka Izbo! Klub Koalicja Polska kilka miesięcy temu poparł zmiany regulaminu umożliwiające zdalne prowadzenie obrad w okresie, terminie zawitym - do końca bieżącego miesiąca. Nasza zgoda podyktowana była racjonalną zasadą ostrożności. Wówczas nie wiedzieliśmy, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia. Widzieliśmy nieradzącą sobie z dużą liczbą chorych służbę zdrowia we Włoszech. Obecnie słyszymy z ust polityków partii rządzącej, że epidemia jest opanowana. Odmrażamy gospodarkę, wysyłamy ludzi do urn wyborczych, dlatego nie ma powodu, aby politycy byli dalej traktowani jak uprzywilejowana kasta. W tym miejscu należy powiedzieć, iż parlament w trakcie ostatnich miesięcy był traktowany wyjątkowo. Przed obradami Sejmu budynki sejmowe były odkażane, a posłowie mieli mierzoną temperaturę. Takiego traktowania nie doświadczyły miliony Polaków, czego pokłosiem jest tragiczna sytuacja w śląskich kopalniach, a właściwie w całym województwie. Obecnie Sejm pracuje w formie szczątkowej. Nie pracują zespoły parlamentarne, na posiedzenia komisji nie jest wpuszczana strona społeczna, a same posiedzenia komisji są zwoływane sporadycznie. Przedstawię konkretny przykład. Jeśli chodzi o komisję rolnictwa, to do dnia dzisiejszego odbyło się 15 posiedzeń, a w ubiegłej kadencji w identycznym okresie odbyło się 50 posiedzeń, czyli ponad trzy razy więcej. Reasumując, nie wyrażamy zgody na dalsze pozorowanie prac Sejmu, dlatego składam wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I stanowisko Koła Poselskiego Konfederacja w pierwszej kolejności przedstawi pan poseł Krystian Kamiński. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Rozmawiamy dzisiaj o projekcie, który ma przedłużyć działanie nowego regulaminu Sejmu. Dlaczego w momencie odmrażania gospodarki, uspokajania obywateli i wracania do normalnego życia posłowie mają być inaczej traktowani i nie muszą wracać do normalnego trybu pracy? Odpowiedź jest prosta: ponieważ Prawu i Sprawiedliwości taki sposób zdalnego procedowania jest na rękę. Wszyscy wiemy, że nie jesteście w stanie upilnować swoich posłów, którym nie chce się przyjeżdżać na posiedzenia Sejmu, którym nie chce się przyjeżdżać na posiedzenia poszczególnych komisji, którym odpowiada to, że wystarczy zalogować się do systemu, kliknąć w ikonkę i pełna wypłata wpłynie na konto. Nawet nie muszą oni oglądać obrad Sejmu czy komisji. Tylko czy tak ma wyglądać praca polskich parlamentarzystów? Zdaniem Konfederacji zdecydowanie nie. W ostatnim czasie mieliśmy rozmawiać o kilku umowach międzynarodowych oraz opiniować przyszłych polskich ambasadorów. Na 29 posłów w posiedzeniach komisji na miejscu brało udział 4, w porywach do 7 posłów. System Polycom, dzięki któremu posłowie teoretycznie mogą brać udział zdalnie w posiedzeniach, działa wybiórczo.

Czy tak ma wyglądać poważna debata nad bardzo istotnymi tematami? To jest kpina z parlamentaryzmu, ale również z Polaków, ponieważ w ich interesie powinniśmy pracować, a nie siedzieć w domu. Dodatkowo uniemożliwia się udział w komisjach stronie społecznej i ekspertom w danych dziedzinach, co prowadzi do zaniżenia poziomu debaty. Obecne brzmienie regulaminu służy pani marszałek do ograniczania czasu wypowiedzi z mównicy. Drastycznym tego przykładem było przeznaczenie zaledwie kilku minut na przedstawienie obywatelskich projektów ustaw o ochronie życia poczętego bądź przeciwko ustawie 447, pod którymi podpisały się setki tysięcy, a nawet miliony Polaków. Odrzućmy to wygodnictwo zdalnego udziału w posiedzeniach, reglamentacji Sejmu i wróćmy do normalnej pracy, prowadząc normalną debatę dla dobra wszystkich Polaków. Przechodzimy do pytań. Przechodzimy do pytań. Wyznaczam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Zamykam listę. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Mam pytanie do pani poseł wnioskodawcy. Jaki miernik epidemii sugeruje utrzymanie zdalnych posiedzeń Sejmu? Tak jak napisaliście państwo w projekcie uchwały, chcecie, aby utrzymało się bezterminowo zdalne posiedzenie Sejmu, dlatego że obowiązuje stan epidemii. Mowa o stanie epidemii, o którym nasz dzielny premier Morawiecki i dzielny minister Szumowski mówią, że go nie ma, krzywa się wypłaszczyła. Odmrożono galerie handlowe, odmrożono bardzo wiele dziedzin życia społecznego i gospodarczego, wpuszczono tam Polaków. Chcemy pracować normalnie, tak jak pracują wszyscy Polacy. My chcemy pracować normalnie i rzetelnie. Dlaczego chcecie, żeby były zdalne posiedzenia? Bo nie chcecie, żeby opozycja miała głos, żeby opozycja była aktywna. Dziękuję bardzo.

Panowie Posłowie! Biorąc pod uwagę ciągle rozwijającą się epidemię koronawirusa w Polsce i nieporadność rządzących w jej zwalczaniu, nie dziwi umożliwienie zdalnych posiedzeń Sejmu, ale, proszę państwa, to nie jest uzasadnienie dla zwoływania posiedzeń komisji przez marszałek, a nie przez poszczególnych przewodniczących. Jak pokazały ostatnie 4 miesiące, taki zapis praktycznie blokuje rzetelną pracę nad ustawami. Wczorajszy przykład - Komisja Polityki Senioralnej zebrała się po raz pierwszy od połowy lutego wczoraj, na 15 minut. Nikogo nie obchodzą zakażenia w DPS-ach, trudna sytuacja seniorów. 15 minut poświęcono wczoraj na obrady Komisji Polityki Senioralnej. Nie chcę już nic mówić o tym, że jeśli nie ma posiedzeń komisji, nie mogą głosu zabrać także osoby, które pracują w organizacjach społecznych. Te rozwiązania nie usprawniają pracy komisji, tylko ją marginalizują, a chyba nie o to nam chodzi. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dobromir Sośnierz, koło Konfederacja. Bardzo proszę. Nie rozumiem, dlaczego robimy ten wyjątek dla naszej Wysokiej Izby.

Prosiłbym o wyjaśnienia.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Ta dzisiejsza nasza niby-debata tak naprawdę potwierdza tylko to, że nigdy nie chodziło o zdalne czy elektroniczne obradowanie, a COVID był tylko pretekstem. Tak naprawdę chodziło i chodzi o to, żebyśmy nie tyle mieli Sejm niemy, ile Sejm na smyczy, nawet jeśli bezprzewodowej, Sejm na pilota sterowanego z Nowogrodzkiej. To też nie osobiście, bo nie sądzę, że szeregowy poseł jest tak cyfrowo zaawansowany. I to jest prawda o tym waszym projekcie, zwłaszcza że przypominamy sobie, nie było to tak dawno, że pierwotnie to miało być rozwiązanie właśnie terminowe. To była umowa dżentelmeńska ze strony opozycji, że zgodzimy się wtedy, kiedy będzie potwierdzenie, że to jest krótkotrwałe. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przyjęte zmiany w zakresie umożliwienia wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość miały swój cel i nie ulega wątpliwości, że było to potrzebne rozwiązanie w momencie wzrostu zakażeń. Ale, proszę państwa, moi wyborcy, jak pewnie i państwa, głosowali na mnie w województwie podlaskim i niczym się nie różnimy od fryzjerek, kosmetyczek, lekarzy. Powinniśmy pracować w miejscu pracy, do czego zostaliśmy wybrani. Lewica jest za tym, żebyśmy pracowali już tylko i wyłącznie w Sejmie. Pan poseł Krzysztof Piątkowski, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Szanowni Państwo! Czyli jak? Czyli marszałek będzie decydował, ile osób, ilu polskich posłów będzie mogło wejść na salę obrad? Ile osób będzie mogło zabrać głos w dyskusji? Szanowni Państwo! O jakie przesłanki chodzi? To państwo dzisiaj decydujecie o kształcie polskiego parlamentu. Wszyscy, którzy dziś zagłosują za tym, powinni mieć świadomość tego, że przejdą do historii jako ci, którzy ograniczyli rolę i znaczenie polskiego parlamentu i sprowadzili tę rolę do roli parlamentu kanapowego, nieistotnego. Ja nie zostałem wybrany na kanapowego posła, tylko na posła, który ma reprezentować w sposób właściwy interes swoich wyborców.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Posłowie! Nie pytajcie się, dlaczego to jest wprowadzone. Nie pytajcie się, dlaczego nie można przyprowadzić do Sejmu ekspertów, dlaczego to marszałek Sejmu odebrał przewodniczącym komisji zdolność zwoływania posiedzeń poszczególnych komisji. Nie pytajcie się o takie szczegóły. Zdajmy sobie sprawę na tej sali z jednej rzeczy: tak jak COVID19 wyniszcza płuca ludzkie w wyniku patogenu, tak Zjednoczona Prawica pod sztandarami Jarosława Kaczyńskiego wyniszcza płuca demokracji, jakimi jest parlament. To jest istota tego zabiegu.

Wysoka Izbo!

Do mnie pani mówi? Ja przeczytałem.

Jestem w dwóch komisjach.

Dlaczego nie chcecie pozwolić, żebyśmy mogli normalnie pracować (Dzwonek), żebyśmy mogli procedować nad tym, czego ludzie od nas oczekują? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szeregowy Pośle Kaczyński! Wysoka Izbo! Przychodząc do Sejmu, naiwnie miałam nadzieję na to, że zobaczę tu prawdziwy parlamentaryzm, bo przecież samo słowo pochodzi od francuskiego słowa „parler”: mówić, rozmawiać. Jeżeli po coś powinniśmy siedzieć tutaj do nocy, to nie po to, żeby wasze ustawy przechodziły w 1 dzień bez konsultacji społecznych, ale właśnie po to, by dyskutować do woli, by w wyniku tych dyskusji ustanawiane było jak najlepsze prawo. W zamian tego, pod przykrywką pandemii i z powodu wątpliwej jakości głosowania zdalnego, zobaczyłam zupełne tego zaprzeczenie. Będzie pytanie, mam czas. Partia rządząca wykorzystała epidemię, by nawet Sejm sprowadzić do jego parodii: cicho, szybko, bez mediów, a posłanki i posłowie zostali sprowadzeni do zdalnych maszynek do głosowania. Czy naprawdę chcemy ten stan, zdalny Sejm niemy przedłużyć. Dziękuję. Było pytanie. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Obecny parlament, działający na podstawie regulaminu, którego obowiązywanie chcecie państwo przedłużyć, to fasada parlamentaryzmu. Dyskusje nad projektami są żałośnie fasadowe. Pani marszałek redukuje debaty do 3 minut i trzech pytań na klub. Pani marszałek non stop obchodzi regulamin, skracając do zera czas na zapoznanie się z projektami. Posiedzenia komisji są fasadowe, od marca praktycznie się nie odbywają. Komisja wodna nie zajęła się planem „Stop suszy!”, komisja energii nie zajmuje się dramatyczną sytuacją w kopalniach, członkowie komisji odpowiedzialnej za klimat na oczy nie widzieli ministra klimatu. Może ktoś go widział? A przecież posiedzenia zdalne teoretycznie mają umożliwić i dyskusję, i same posiedzenia komisji. Dlaczego one się nie odbywają? Czy przedłużając trwanie, obowiązywanie tego regulaminu w nieskończoność chcecie państwo w nieskończoność przedłużać fasadowość polskiego parlamentaryzmu? Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam dość. Mam tak samo demokratyczny mandat jak każdy inny poseł z PiS-u. Zostałam wybrana głosami moich wyborców i powinnam mój mandat realizować w sposób niezawisły, demokratyczny i niczym nieograniczony. Tymczasem państwo mi go bardzo ograniczacie. Mało tego, państwo jeszcze nam skracacie czas zadawania pytań i do tego, proszę państwa, przerywacie nie tylko w połowie zdania, lecz również czasami nawet w połowie słowa. Chcę realizować swój mandat poselski tak jak każdy inny poseł. Parlament nie może być zamknięty dla posłów. Parlament jest właśnie po to, żebyśmy tutaj się spotykali, ścierali podczas dyskusji i tworzyli dobre prawo. Jak mamy się spotykać, skoro jesteśmy [[Dzwonek]] aktywni tylko w Internecie? Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę. Mamy dość ograniczania posłom możliwości wykonywania normalnej pracy. Mamy dość blokowania dostępu do sali plenarnej. Mamy dość blokowania posiedzeń komisji. Mamy dość braku możliwości pracy zespołów. Mamy dość ograniczania wystąpień posłów w Sejmie. Mamy dość blokowania udziału strony społecznej w pracach parlamentu. I mamy dość ograniczania dyskusji nad przepisami, które dotyczą wszystkich Polaków. Mamy dość tego reżimu, który niszczy polski parlamentaryzm. I mam jedno pytanie: Czy wy w PiS-ie nie widzicie, że Polacy też mają tego wszystkiego serdecznie dość?

Czym w praktyce jest zdalny Sejm? Niczym innym jak ograniczaniem naszych praw, które dali nam wyborcy, wybierając nas do parlamentu. Jak wygląda zdalna praca Sejmu? Tak naprawdę jestem posłem Komisji Finansów Publicznych, która w czasie epidemii pracuje non stop, zbiera się praktycznie co tydzień, bo stała się specjalistą już nie tylko od prawa dotyczącego finansów publicznych, ale również nawet od Kodeksu karnego. I jak wygląda praca w tej komisji? Posłowie siedzę przed swoimi tabletami z takimi karteczkami: proszę o głos - Paulina Hennig-Kloska. Czy jest nam udzielany głos? Czy możemy dowolnie składać poprawki, chcąc stanowić dobre prawo? Nie, bo najzwyczajniej jest to tylko i wyłącznie dobra wola przewodniczącego i posłowie Prawa i Sprawiedliwości za każdym razem ten głos dostają, a posłowie opozycji - nie. Mamy dość reżimu parlamentarnego, [[Dzwonek]] który tutaj wprowadziliście, który nie ma nic wspólnego z dobrym stanowieniem prawa i z dbaniem o prawa i wolności obywateli. Dziękuję bardzo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Zamykam. Aha, o głos prosiła pani poseł Barbara Bartuś. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Trochę logiki w tym wszystkim. Kilkudziesięciu posłów z mównicy krzyczało, że nie może zabrać głosu. Nie było pytań.

Bardzo proszę. Było dość czasu, żeby się z nimi zapoznać. Szanowni państwo, te przepisy stanowią, że Sejm w trybie zdalnym może - może, nie musi, ale może - być tylko wtedy zwołany, kiedy mamy stan epidemii lub jeden z trzech stanów nadzwyczajnych, które są wymienione w konstytucji. I nie ma takiej możliwości, aby w innym czasie, bez stanu klęski żywiołowej czy bez stanu epidemii, tych przepisów użyć. Decyduje marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Tak, bo marszałek organizuje prace Sejmu.

Pozwólcie, że odpowiem wam na pytania, ponieważ tak naprawdę było to krzyczenie tylko po to, żeby pokrzyczeć, natomiast nie rozumiecie, że jeżeli chodzi o. możliwość dostępu do pracy, to te przepisy na to pozwalają. Szanowni Państwo! Gdy była sytuacja bardzo trudna, były ograniczenia tutaj, na sali sejmowej, tak żeby było mniej osób. Wtedy były ograniczenia i były też zapewnione sale komisyjne, tak że każdy poseł, który chciał, mógł przyjechać, mógł brać udział w posiedzeniu. W tej chwili, skoro sytuacja w Polsce się poprawiła. to wiecie państwo, że wchodzi każdy poseł, który chce wejść. Szanowni Państwo! Jednak jesteście na tej sali. A do pani poseł Jachiry: pamiętam taki filmik, kiedy pani się naigrywała, jaki to Sejm polski jest zacofany, że nie można elektronicznie. To niech pani się zdecyduje, czy pani chce elektronicznego głosowania, czy nie.

To dzięki temu, że mieliśmy takie rozwiązania, mogliśmy tak procedować. Jeszcze raz podkreślę: ten artykuł dotyczy zniesienia.

Dlatego prosimy o to, żeby po prostu skreślić ograniczenie czasowe, zostawić to w regulaminie po to, żeby, jeżeli kiedyś byłaby taka sama sytuacja, jak nas spotkała w tym roku, takie przepisy móc. Szanowni Państwo! Stan epidemii... zachorowania się wypłaszczyły. To nie znaczy, że nie może się tak zdarzyć, że ktoś z państwa za tydzień będzie w kwarantannie i nie będzie mógł przyjechać na posiedzenie Sejmu.

I tak samo ministrowie, nasi posłowie w sytuacji bycia w kwarantannie mogli nie być wyłączeni z możliwości brania udziału w posiedzeniach, głosowaniach, a to jest nasze prawo. Konfederacja powiedziała, że komuś się nie chce. A Konfederacja to jest chyba ten klub. Zadawali pytanie, Konfederacja zadawała pytanie, więc odpowiadam. Dlatego też jeszcze raz, szanowni państwo, proszę o przemyślenie. Nie można tych przepisów zastosować w innej sytuacji.

I jeżeli stan epidemii się zakończy. te przepisy nie będą mogły być używane, ale jeżeli za rok, za 2, za 5 lat stałoby się tak, że jakiś stan nadzwyczajny zostanie ogłoszony, mielibyśmy gotowe przepisy, nie musielibyśmy wtedy myśleć, jak ma obradować Sejm. Dlatego jeszcze raz państwa proszę. Dla nas wszystkich, dla nas, parlamentarzystów, którzy chcą pracować, jest to dobre rozwiązanie.

Panie posłanki, jeśli chcecie jeszcze porozmawiać, to zawsze jest okazja w kuluarach, dobrze? W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu uchwały oraz o przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania. Do głosowania nad tymi wnioskami przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 388) Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana Rafała Webera o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę, panie ministrze.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić projekt zmian bardzo długo oczekiwanych przez właścicieli pojazdów samochodowych, projekt zmian, które z jednej strony przyczynią się do likwidacji pewnych obowiązków administracyjnych, ale z drugiej strony przyczynią się również do likwidacji pewnych obowiązków związanych z opłatami, z finansami, które w tej chwili są obowiązkowym elementem, kosztem poniesionym przez właścicieli pojazdów samochodowych. Szanowni Państwo! Na wstępie tego swojego wystąpienia chcę bardzo gorąco podziękować w imieniu pana ministra Andrzeja Adamczyka wszystkim tym, którzy współpracowali z resortem infrastruktury przy tworzeniu tego pakietu zmian. Bardzo gorąco dziękuję panu ministrowi Markowi Zagórskiemu, ministrowi cyfryzacji oraz całemu zespołowi Ministerstwa Cyfryzacji, który też swoim wkładem, swoją chęcią zmian w tym zakresie przyczynił się do powstania tego projektu ustawy. Bardzo gorąco dziękuję również ministrowi spraw wewnętrznych i administracji panu Mariuszowi Kamińskiemu, wiceministrowi panu Pawłowi Szefernakerowi, ponieważ właśnie w tym trójkącie resortów ustalaliśmy te najważniejsze rzeczy, najważniejsze kwestie związane z tym projektem. Drodzy Państwo! Zostały mi 3 minuty 30 sekund na to, aby przedstawić najważniejsze założenia tego projektu. Oczywiście nie uczynię tego, bo tego czasu jest za mało. Oczywiście jesteśmy do państwa dyspozycji, jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania, które pojawią się za chwileczkę zarówno w wystąpieniach klubowych, jak i w wypowiedziach poszczególnych posłów. Natomiast bardzo krótko o tych najważniejszych zmianach, o tych najważniejszych korzyściach dla właścicieli pojazdów w Polsce. Drodzy Państwo! Likwidujemy obowiązek posiadania karty pojazdu, likwidujemy obowiązek posiadania nalepki, pozwalamy na to, aby stare tablice rejestracyjne mogły być niezmieniane, mogły być przypisywane do właściciela, który rejestruje samochód w Polsce, tak aby ten numer rejestracyjny cały czas mógł iść za nim. Jest to oczywiście związane z ułatwieniem administracyjnym, ale także z brakiem opłat, które są związane z wymianą tablic rejestracyjnych. Kolejna zmiana, bardzo istotna: prawo jazdy zostaje w domu. Nie będzie obowiązku posiadania przy sobie, kierując samochodem, prawa jazdy i okazywania go w trakcie kontroli drogowej. W razie kontroli czy to policjant, czy to inspektor Inspekcji Transportu Drogowego będzie mógł w systemie odszukać, czy faktycznie osoba kierująca pojazdem posiada uprawnienia do tego, aby kierować pojazdem, czy to do 3,5 t, czy to później pojazdem ciężkim. Umożliwiamy czasową rejestrację w miejscu zakupu samochodu. Nowy właściciel pojazdu będzie miał możliwość czasowej rejestracji pojazdu przez organ rejestrujący właściwy dla miejsca zakupu pojazdu. Dzięki temu w przypadku konieczności przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu oraz... lub odbioru do miejsca zamieszkania nowy właściciel zarejestruje czasowo pojazd u miejscowego, czyli u tego, u którego sobie ustali, wybierze, starosty. Nie będzie już musiał jeździć do miejsca zamieszkania, aby czasowo zarejestrować samochód kupiony w innej części kraju. Kolejny ważny element: uporządkowanie rejestracji wywożonych pojazdów w przypadku wydania pozwolenia czasowego na wywóz pojazdu za granice Polski i złożenia przez właściciela pojazdu oświadczenia, że pojazd zostanie wywieziony, organ wyrejestruje ten pojazd z urzędu. To pozwoli uporządkować sytuacje, kiedy samochód jest sprzedawany poza granice kraju. Następny element: rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z eksploatacji o samochody osobowe. Kolejny element: właściciel pojazdu, zmieniając miejsce zamieszkania na terytorium Polski, nie będzie musiał przedstawiać dowodu własności pojazdu, przerejestrowując swój samochód u innego starosty. Do wniosku o rejestrację wystarczy dowód rejestracyjny z aktualnymi (Dzwonek) badaniami technicznymi i nie będzie potrzeby dostarczać do urzędu umowy kupna pojazdu. Po wygaśnięciu ważności czasowych pozwoleń właściciel nie będzie musiał zwracać nieważnych już dokumentów do urzędu. Jedenasta zmiana: diler będzie mógł sam zarejestrować nowy samochód w trybie online. Kolejna zmiana - i tutaj usługa Ministerstwa Cyfryzacji - tzw. „Mój pojazd”, czyli umożliwienie generowania i wydruku raportu z udostępnianej przez ministra cyfryzacji usługi „Mój pojazd” i nadanie temu wydrukowi mocy dokumentu potwierdzającego dane zgromadzone w centralnej ewidencji pojazdów. I zmiana jeszcze jedna - dowód rejestracyjny bez miejsca na stemple też będzie cały czas w obrocie. Szereg bardzo potrzebnych, bardzo istotnych zmian, ułatwień administracyjnych, odciążeń finansowych. Mam nadzieję, że Wysoka Izba w całości poprze ten projekt zmian i razem z nami, razem z rządem Prawa i Sprawiedliwości, z Ministerstwem Infrastruktury, wdroży te nowe przepisy do polskiego porządku prawnego. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Piotr Król. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko co do projektu ustawy o zmianie Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 388. Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg ułatwień dla obywateli, w tym zarówno właścicieli pojazdów, jak i przedsiębiorców, oraz zmniejsza w związku z tym odpowiednio zakres zadań i obciążenia administracyjne organów samorządowych. Wśród najistotniejszych propozycji zainicjowanych przez ministra infrastruktury znajdują się następujące regulacje realizujące oczekiwania społeczne. Po pierwsze, projekt umożliwia zachowanie na wniosek właściciela pojazdu dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, jeżeli właściciel pojazdu składa wniosek o rejestrację pojazdu, który był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po drugie, znosi obowiązek wydawania karty pojazdu w procesie pierwszej rejestracji pojazdu. Po trzecie, znosi obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeśli od uprzedniej, ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie własności pojazdu. Przewidziano również propozycję umożliwienia czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku konieczności przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu. Z kolejnych ułatwień, o których warto wspomnieć, najistotniejsze jest zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dokumentu prawa jazdy. Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw możliwości nieposiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego. Poza tym umożliwia się rejestrację drogą elektroniczną nowego pojazdu samochodowego przez przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą nowych pojazdów samochodowych w imieniu kupującego. Znosi się również obowiązek wydawania tzw. nalepki kontrolnej. Ponadto w projekcie ustawy zawarto również inne zmiany regulujące na poziomie ustawy obecne rozwiązania systemowe poprawiające legalność obrotu pojazdami i referencyjność danych gromadzonych w CEPiK. W związku z tymi zmianami w ustawie Prawo o ruchu drogowym przewidziano również zmiany w innych ustawach, np. w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawie o kierujących pojazdami czy ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Klub Prawa i Sprawiedliwości zamierza aktywnie wspierać uchwalenie tego projektu. Dziękuję bardzo, panie pośle. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Franciszek Sterczewski. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Zaproponowane przez rząd rozwiązania przedstawione w ramach czytanej dzisiaj zmiany Prawo o ruchu drogowym spowodować mogą nie tylko dodatkowe problemy dla kierowców, ale także dla urzędów, które zajmują się rejestracją pojazdów. Od wielu lat rozmawiamy o cyfryzacji urzędów, która pomogłaby w załatwianiu wielu codziennych spraw. Ostatnie miesiące, czas epidemii, pokazały, jak potrzebne może być przeniesienie procedur do świata wirtualnego. Problem tkwi w tym, że cyfryzacja powinna być wprowadzana w sposób przemyślany i spójny, w przeciwnym razie może przynieść więcej szkód niż pożytku. Doskonale pamiętamy, jaki chaos w urzędach spowodowało wprowadzenie jesienią 2017 r. systemu CEPiK 2.0. W całej Polsce wydziały komunikacyjne zostały sparaliżowane, a petenci tkwili w długich kolejkach. Proponowany projekt ustawy może być powtórką z tej wątpliwej rozrywki. Na pierwszy rzut oka ustawa wprowadza kilka ułatwień: likwiduje kartę pojazdu, naklejkę kontrolną oraz wprowadza możliwość zachowania tablic rejestracyjnych przy przerejestrowywaniu pojazdu. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Pod wieloma względami uciążliwa procedura rejestracji pojazdu pozostanie niezmieniona. Zdecydowanej większości spraw wciąż nie będzie można załatwić od A do Z przez Internet, a wiele zbędnych formalności pozostanie.

Autorzy projektu informują, że wprowadzone rozwiązania znacznie zmniejszą zakres zadań organów rejestrujących pojazdy. To jednak nieprawda, o czym wyraźnie mówią przedstawiciele samorządów. Rozmawiałem z urzędnikami z Wielkopolski. Ostrzegali, że proponowana ustawa może jeszcze bardziej skomplikować ich pracę, ponieważ rozwiązania nie są ze sobą spójne, a poszczególne systemy nie współpracują ze sobą. Także Związek Powiatów Polskich w skierowanym w lutym br. liście do premiera Mateusza Morawieckiego wzywał do zawieszenia prac nad tą ustawą i ostrzegał przed chaosem w systemie rejestracji pojazdów. Urzędników i urzędniczki czeka ta sama praca, wciąż będą musieli przeprowadzać podobne postępowanie administracyjne i wydawać decyzje o rejestracji pojazdu. Dodatkowo powierzone im zostaną nowe zadania, takie jak chociażby ocena zdatności odnośnie do rejestracji tablic. Dlaczego proponowane są przepisy, które z perspektywy urzędów generują jeszcze większy chaos? Równocześnie ograniczony zostanie dochód jednostek samorządu terytorialnego. Dla wielu mniejszych samorządów może to być poważny problem. Przed tym także ostrzega Związek Powiatów Polskich. To oznacza ograniczenie liczby etatów i w praktyce dłuższe kolejki w wydziałach komunikacji. Ograniczenie dochodów samorządowych jest niestety zgodne z polityką rządu, która rzuca polskim miastom kłody pod nogi. To budzi mój zdecydowany sprzeciw. Dlatego mam kolejne pytanie: Jak rząd planuje zrównoważyć ubytek dochodów samorządów? Obecny system jest niespójny, wymaga prawdziwej reformy. Kierowcy i urzędnicy zasługują na stworzenie kompletnego rozwiązania, umożliwiającego realizowanie formalności od początku do końca za pomocą jednego systemu. Ustawa w tej formie nie staje na wysokości zadania.

Czy to oznacza, że ta ustawa jest tylko próbą przypodobania się kierowcom w czasie kampanii prezydenckiej, a tak naprawdę jej wejście w życie chcecie przekładać na święte nigdy? Ta ustawa wymaga bardzo istotnych zmian, dlatego klub Koalicji Obywatelskiej jest za skierowaniem jej do dalszych prac w komisji. ale pod warunkiem, że dalsze prace będą oparte na dialogu z samorządami, stroną społeczną i ekspertami. Nie zgadzamy się, by prawo było tylko zasłoną dymną, która teoretycznie niektóre kwestie rozwiązuje, a z drugiej strony utrudnia życie kierowców i urzędów. Dziękuję bardzo, panie pośle. I pani poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ze stanowiskiem klubu Lewica. Bardzo proszę, zapraszam panią poseł. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Uproszczenie warunków i trybów rejestracji pojazdów to naszym zdaniem słuszne działanie, odpowiednio wdrożone może przełożyć się na odciążenie urzędów i ułatwienie życia obywateli i obywatelek. Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie i okazywania prawa jazdy podczas kontroli, posiadania nalepki kontrolnej z numerem rejestracyjnym czy też wprowadzenie możliwości pozostawienia dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy jego przerejestrowaniu to zdaniem Lewicy sensowne i ułatwiające życie działanie. Dlatego Lewica zagłosuje za dalszymi pracami nad prezentowanym projektem ustawy. Ale omawiając zmiany w Prawie o ruchu drogowym nie sposób nie przypomnieć o tych, na które naprawdę czekają miliony Polek i Polaków. Każdego roku na polskich drogach ginie ok. 3 tys. osób, ponad 35 tys. traci w zdarzeniach drogowych zdrowie. Nie mam wątpliwości, że rząd premiera Morawieckiego jest w pełni świadomy tych smutnych danych. Jest świadomy na tyle, że w listopadowym exposé pan premier bezpieczeństwo ruchu drogowego odmieniał przez wszystkie przypadki i obiecywał istotne zmiany chroniące pieszych i innych słabszych uczestników ruchu drogowego. Te obiecywane zmiany to nie tylko zmiany istotne, ale co ważne, bardzo łatwe i proste do szybkiego wdrożenia. Realne pierwszeństwo pieszych na pasach, ujednolicenie limitów prędkości w terenie zabudowanym, zaostrzenie kar dla bandytów drogowych i odbieranie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km/h czy w końcu przebudowa miejsc niebezpiecznych - to naprawdę proste zmiany. Zwłoka w ich wdrażaniu to odmowa ratowania życia tysięcy Polek i Polaków. I o ile ułatwienia procedur rejestracyjnych dla kierowców są sensowne i być może potrzebne, o tyle tak naprawdę to ochrona życia i zdrowia powinna być najwyższym priorytetem rządu. Przez brak obiecanych przez premiera zmian w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego polskie drogi są wciąż jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Unii Europejskiej, a w rankingu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Polska spadła na trzecie miejsce od końca. Dziś więcej ludzi ginie już tylko na drogach w Bułgarii i w Rumunii. To powinno być wielkim wyrzutem sumienia obecnego rządu, bo pokazuje, że pan premier Morawiecki i rząd Prawa i Sprawiedliwości, podobnie jak rząd poprzedniej ekipy, nie uznaje tych koniecznych dla ochrony życia zmian za priorytet. Do przyspieszenia prac w tym zakresie nie mobilizuje rządu smutna rzeczywistość polskich dróg i regularne informacje o tragediach spowodowanych przez bandytów drogowych ignorujących ograniczenia prędkości czy prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu. Niestety wciąż nie słychać też o programie inwestycji przebudowy miejsc niebezpiecznych, mimo że taka inicjatywa mogłaby być ważnym elementem planu naprawy życia społecznego i gospodarczego po kryzysie spowodowanym epidemią koronawirusa. Wysoka Izbo! Przedłożony przez rząd projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym nie jest, zdaniem Lewicy, projektem złym. Nasze wątpliwości budzi jednak fakt, że dla obecnego rządu kwestia rejestracji pojazdów ważniejsza jest od ludzkiego życia. W imieniu swoim i Lewicy apeluję do pana premiera, do ministra infrastruktury i do rządu o jak najszybsze procedowanie nad kluczowymi zmianami w Prawie o ruchu drogowym, tymi zmianami, na które naprawdę wszyscy czekamy.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 388. Czytamy, że celem nowelizacji ustawy są uproszczenia w kontekście oczekiwań społecznych, jeśli chodzi o zmniejszenie kosztów i obciążeń administracyjnych dla posiadaczy pojazdów. W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie rozwiązań, które można by pogrupować.

I tutaj już do tej zmiany odniósł się Związek Powiatów Polskich, który powiedział, że projekt w przedłożonym kształcie nie był opiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, co stanowi naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Równocześnie należy dodać, że poprzednia wersja projektu została negatywnie zaopiniowana przez Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Trudno mówić o tym, że to będzie zmniejszona ilość zadań dla organów rejestrujących pojazdy, skoro jak już wcześniej wskazywano, organ będzie musiał oceniać zgodność tablic rejestracyjnych, będzie także musiał wykonywać czynności związane z rejestracją tych pojazdów. Będą oczywiście obywatele zmuszeni i tak dwukrotnie udać się do urzędu. Znając życie, to i tak urzędnicy będą prosić o te dane i właściwe dokumenty. To jest tak jak z e-dowodem, który wszędzie ma działać. Okazuje się, że w urzędach, w bankach jesteśmy proszeni, żeby jednak wyjąć z kieszeni dowód i fizycznie go okazać. To jest tak jak w polskiej komedii „Kogel-mogel”: łazienka jest, bo co by powiedzieli, że u nas łazienki nie ma?

Tu chociażby StowarzyszenieKomisów.pl mówi o tym, żeby udostępnić możliwość rejestracji pojazdów przez Internet wszystkim obywatelom i przedsiębiorcom, a nie tylko salonom samochodowym, żeby zastąpić obowiązek rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej obowiązkiem tylko zgłoszenia nabycia pojazdu i umożliwić posługiwanie się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalną tablicą rejestracyjną również w przypadku wykonywania przez podmioty uprawnione jazd próbnych samochodami niezarejestrowanymi wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź samochodami osobowymi przeznaczonymi do sprzedaży i wycofanymi czasowo z ruchu. Dlatego też ważne jest, żeby każdy z Polaków miał możliwość chociażby wyrejestrowania auta, zawieszenia na jakiś czas, niepłacenia ubezpieczenia, kiedy z tego auta nie korzysta.

Oby tak się stało, będziemy temu kibicować. Stanowisko Koła Poselskiego Konfederacja przedstawi pan poseł Dobromir Sośnierz. Bardzo proszę. To chyba będzie pierwsza w tej kadencji większa ustawa, którą będę mógł tutaj z czystym sumieniem pochwalić. Próbowałem w niej znaleźć jakieś tam haczyki i niebezpieczeństwa, bo przyzwyczailiście nas państwo już do tego, że każdy wasz przepis trzeba oglądać pod światło dziesięć razy i zastanawiać się, co tam zachachmęciliście w tym, no ale na razie nie znalazłem nic złego. Nie gasimy czujności, ale na razie plus dla was. Jak zobaczyłem ten tytuł w porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, to już, szczerze mówiąc, spodziewałem się najgorszego, że ministerstwo w samobójczym jakimś odruchu tuż przed wyborami odgrzebało ten zapowiadany wcześniej głośno i tutaj przypominany już, ale naprawdę głupi i szkodliwy pomysł kolejnych zmian przepisów dotyczących porządku przechodzenia przez jezdnię i ograniczeń dla kierowców. Na szczęście przed wyborami PiS schował kij za plecami i macha marcheweczką, taką tam niedużą, ale jednak zawsze, więc doceniam. Uproszczenie procedur, rezygnację z archaicznych wymagań dotyczących okazywania oryginalnych dokumentów oraz posiadania przy sobie dokumentów, które bez trudu może sobie każdy policjant sprawdzić w bazie danych, co daje mu zresztą przecież dużo większą pewność niż oglądanie kawałka plastiku, który łatwiej podrobić niż wpis w centralnej bazie. 20 lat za późno, ale nie wybrzydzajmy.

Nareszcie, nareszcie. Szkoda, że o ile w takich różnych złych i szkodliwych projektach jesteście wręcz zuchwale odważni czasami, to w takich sprawach słusznych postępujecie nieśmiało jak pensjonarka i tak po kawałeczku ograniczacie możliwość wyrejestrowania auta tylko do 12 miesięcy, obarczacie różnymi zastrzeżeniami. Od razu unosi się tam nad tymi przepisami swąd lekkiego lobbingu ze strony zakładów złomujących i stacji kontroli pojazdów, co zresztą tam w uzasadnieniu jest w oszczędnych, ale dość jasnych słowach powiedziane, że bierzemy pod uwagę tutaj interesy tych, którzy mają zarobić na tych przepisach.

Ale mam nadzieję, że nie ulegniecie państwo tym bałamutnym argumentom, które tam są podnoszone, i konsekwentnie, także po wyborach, będziecie stali po stronie obywateli bezlitośnie wyzyskiwanych przez te dotychczas absurdalne przepisy, kiedy trzeba ubezpieczać auto stojące gdzieś na cegłach w warsztacie. Ja sam miałem przypadek, że przez rok nie mogłem korzystać z samochodu, a cała składka roczna OC przeleciała, a więc rozumiem ten ból. Te lękliwe przepisy nie likwidują niestety wielu problemów. Człowiek, który chciałby przerobić samochód na dekorację w ogródku albo trzymać pozbawioną kół przyczepę na działce jako domek dla dzieci, nadal nie będzie mógł tego zrobić bez klękania przed urzędnikami de facto, bo to są urzędnicy, ze stacji złomujących. Na otarcie łez gwarantujecie stacjom kontroli pojazdów dodatkowe badanie techniczne przed ponowną rejestracją. Można się ubiegać o to, żeby je pozostawić.

Widocznie w gonitwie przedwyborczych pomysłów nie starczyło czasu, żeby to doprowadzić do końca.

I w pozostałym czasie koła Konfederacja pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Bardzo proszę. Z przerażeniem zabieram głos, bo przywykłem, że jak coś popieram, to to przepada, a jak coś potępię, to to przechodzi, więc z przerażeniem to popieram. Być może rzeczywiście chodzi tylko o marchewkę przed wyborami, a potem się okaże, że to nieprawda. Ale byłaby to dobra jaskółka. Proszę spróbować złożyć podanie w sądzie, a przekonacie się państwo, że Sejm jest całkowicie otwarty w porównaniu z sądami. Sądy to się dopiero obwarowały przed ludźmi. Dziękuję bardzo, panie pośle. Przechodzimy do pytań. Zamykam listę. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wczytując się w projekt ustawy dotyczącej zmiany przepisów, jeśli chodzi o rejestrację samochodów, dochodzę do wniosku, że w Polsce będzie to przełomowe wydarzenie w tej dziedzinie. Dlatego mam pytanie. Czy według propozycji Ministerstwa Infrastruktury i rządu osoba kupująca nowy samochód będzie go mogła zarejestrować online w salonie samochodowym, w którym to auto nabyła, bez zbędnego jeżdżenia i marnowania czasu na stanie w kolejkach w wydziałach komunikacji urzędów powiatowych czy urzędów miast? Oraz mam drugie pytanie. Chciałbym również zapytać: Czy będzie możliwe, aby osoba kupująca używany samochód mogła sobie zostawić tablice rejestracyjne, na które zarejestrowany był samochód przez poprzedniego właściciela, i po zarejestrowaniu auta mogła nadal z tych tablic korzystać? Dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Natomiast, panie ministrze, mam pytanie dotyczące takiej sytuacji. Otóż w Polsce w bazie centralnej ewidencji pojazdów jest mnóstwo - prawdopodobnie setki tysięcy, jeżeli nie miliony - takich pojazdów, które nie istnieją. One są przypisane do konkretnego obywatela, zarejestrowane i teoretycznie ten obywatel jest w posiadaniu takiego pojazdu, natomiast wszyscy wiemy, że to jest jedno wielkie złudzenie. Te pojazdy nie istnieją z różnych względów, nawet często fizycznie. I pytanie, czy ministerstwo prowadzi prace, bo to by była dobra okazja do unormowania również takiej sytuacji, czyli możliwości pewnego zgłoszenia i wyczyszczenia państwowych baz danych, które (Dzwonek) zawierają nieprawdziwe rekordy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dlaczego w Polsce użytkownik nie może zadeklarować bez potrzeby wyrejestrowywania, że np. od września do maja nie użytkuje pojazdu, który jest wycofany z ruchu? Jest cała masa pojazdów wymagających rejestracji, przeglądów oraz ubezpieczeń, które używane są sezonowo: pługów, ratraków, kamperów i setki pojazdów kolekcjonerskich, które są odstawiane od jesieni do garażu i wyciągane dopiero późną wiosną lub latem. Kolejna kwestia jest otóż taka. Jeśli chodzi o dopuszczalną masę całkowitą pojazdu z przyczepą, to u nas w Polsce przepisy te sięgają jakieś 30 lat do tyłu, [[Oklaski]] czasów, gdy nie istniały jeszcze systemy wspomagania jazdy, hamowania itd. W dzisiejszych czasach żaden właściciel średniej wielkości SUV-a niemający kategorii C nie może wyjechać na drogę, bo są tam przepisy, że może ciągnąć przyczepę o ciężarze nie większym niż 750 kg, czyli przyczepę skonstruowaną dla małego fiata w latach 70. Większość kierowców lekceważy te przepisy, ale my powinniśmy przepisy dostosować do obecnie istniejących realiów, a nie odwrotnie. Bardzo serdecznie dziękuję. ponieważ interesuje to dużą grupę moich wyborców, mógł odpowiedzieć mi na to na piśmie, to będę zobowiązany. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Skoro już założymy, że uda się przeprowadzić te zmiany, to mam takie pytanie: Czy nie warto by było się zastanowić nad tym, żeby część zadań rządowych przekazać samorządom? Skoro zwalniamy moce przerobowe starostw powiatowych, a rząd Prawa i Sprawiedliwości rozbudowuje coraz bardziej aparat władzy centralnej, można by było przekazać pewne zadania powiatom. Na pewno koszt utrzymania jednego etatu i jednego urzędnika w mieście powiatowym jest dużo niższy niż w Warszawie. Skoro ma być łatwiej dla obywateli, skoro ma być lepiej dla samorządów, okej.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Ja mam tylko pytanie do rządu, czy jak tak się już dobrze zaczęło, to nie dałoby się zrobić jakiejś reformy np. w edukacji, bo to jeszcze jest PRL-owska edukacja, czy, powiedzmy sobie, w służbie zdrowia, która jeszcze jest PRL-owska, tam socjalizm działa w najlepsze.

To jest trudniejsza reforma. Widzę, że PiS chce coś zrobić. Liczymy, że również w tych podstawowych dziedzinach też będzie. Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Nie widzę. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Panie Posłanki! Panowie Posłowie! Proponowane zmiany takie jak zniesienie obowiązku noszenia przy sobie prawa jazdy czy zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy jego przerejestrowaniu są zrozumiałe. Jednak przypominam dzisiaj, 19 czerwca, że 1 lipca 2020 r. miały wejść w życie szumnie zapowiadane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i samego premiera Morawieckiego zmiany dotyczące pierwszeństwa w ruchu pieszych oraz wyższych kar dla kierowców. Z tego, co wiadomo, projekt ugrzązł w Ministerstwie Infrastruktury na etapie konsultacji społecznych i nie trafił jeszcze do Sejmu. Przypominam więc rządowi, żeby pochylając się nad poprawą wygody kierowców, nie zapominał o pieszych, którzy bezustannie giną na polskich drogach. Wielu z tych tragedii dałoby się uniknąć, gdybyście wzięli się za regulacje, które obiecywaliście i które są potrzebne. Jeśli to zadanie was przerasta, Lewica chętnie w tym pomoże. Pan poseł Andrzej Szewiński, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nie mam wątpliwości, iż intencją projektodawców było uproszczenie wielu procedur dla właścicieli pojazdów, dla uczestników ruchu drogowego, natomiast często lepsze jest wrogiem dobrego. Chciałbym zaznaczyć, że projekt nie był objęty rzetelnymi konsultacjami społecznymi i nie był przedłożony do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Związek Powiatów Polskich krytycznie również odniósł się do zapisów. Wysoka Izbo! Na samorządy nakłada się obowiązki, pozbawiając źródeł dochodów. I nie jest to też w interesie obywateli. Pomimo niewielkiego zniesienia zadań organów rejestrujących pojawia się pytanie, czy projektodawcy przewidzieli wyrównanie utraconych dochodów dla powiatów, które nie będą w stanie zapewnić odpowiedniej ilości etatów, i w związku z tym wydłuży się czas oczekiwania w wydziałach komunikacji. Dziękuję bardzo. Pan poseł Paweł Krutul, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Super. Prawo jazdy zostaje w domu - superpomysł. Czego jeszcze bym sobie życzył, to już pan minister nie ma na to wpływu - w województwie podlaskim więcej dróg szybkiego ruchu i autostrad. Moje pytanie: Czy rząd rozważa umożliwienie rejestracji pojazdów przez Internet wszystkim obywatelom i przedsiębiorcom, właścicielom pojazdów, również co do samochodów używanych, zamiast ograniczać się do pojazdów nowych? Bardzo proszę o odpowiedź na to. Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof Piątkowski, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Chciałbym poprosić o informację, kiedy rząd spróbuje pomóc samorządom i rozwiązać problem bardzo je dotykający, mianowicie problem związany z coraz bardziej popularnymi, szczególnie w wielkich miastach, elektrycznymi hulajnogami. pędzą chodnikami z prędkością nieraz 65 km/h. Warto byłoby się przez moment zastanowić i uregulować te kwestie. Rozwiązanie jest chyba proste, natomiast trzeba trochę pracy i wysiłku w to włożyć. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.

Panie Ministrze! Po pierwsze, wiemy dobrze, jak działa system CEPiK, jaki miał start i jak to funkcjonuje do dziś czasami z przerwami. I pytanie: Czy brak obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy nie będzie skutkował tym, że obywatele w trakcie kontroli będą musieli długo oczekiwać na weryfikację prawa jazdy w systemie zdalnym, który działa różnie i działa z przerwami? Chciałam zapytać o zdalną rejestrację pojazdów, jak to będzie faktycznie funkcjonowało, ponieważ wydaje się, że aby to poprawiło jakkolwiek sytuację - zwłaszcza w tych powiatach, a ja z takiego pochodzę, gdzie liczba zarejestrowanych pojazdów na mieszkańca jest większa - to system, po pierwsze, musi być względnie spójny, a po drugie, powinien w jakiś sposób być też zdalnie obsługiwany. Czy dalej do wydziałów komunikacji właśnie [[Dzwonek]] w tych niektórych powiatach bardzo przeciążonych, czy będzie to faktycznie zdalnie obsługiwane, tak by rozładować korki w tych najtrudniejszych miejscach? Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę, panie ministrze.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za dyskusję, za pytania, za wypowiedzi. Podzielimy nasze odpowiedzi na dwie części: ja - jedna część, druga część, ta związana z cyfryzacją - pani minister Wanda Buk, która jest obecna z nami na sali plenarnej i której jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję za współpracę przy przygotowaniu tego projektu. Zostawiłem pewną przestrzeń dla państwa, sądząc, że któreś z was podliczy oszczędności finansowe, które dzięki temu projektowi zostaną wygenerowane w kieszeniach Polaków, właścicieli pojazdów, którzy nie będą objęci pewnymi obowiązkami, które w tej chwili są na nich przez nas nałożone czy tam kiedyś zostały nałożone.

W mojej ocenie to bardzo dużo, tym bardziej że w niektórych wypowiedziach posłowie opozycji mówili o uszczupleniu przychodów jednostek samorządu terytorialnego, które w tej chwili zajmują się zadaniami związanymi z komunikacją. Padł nawet przykład, że w ciągu roku jeden z samorządów straci 6 mln zł, czyli, drodzy państwo, 6 mln zł zostanie w kieszeni obywatela. Nie wróci do Skarbu Państwa, nie będzie w dyspozycji ministra infrastruktury czy w dyspozycji ministra finansów, zostanie w kieszeni obywatela. O to chodzi w tym projekcie - oszczędność finansowa i oszczędność czasowa.

Na wszystkie pytania, które tutaj padły, w przypadku których poproszono o odpowiedź pisemną, na pewno taka odpowiedź pisemna zostanie udzielona. Zapraszam państwa do dyskusji na ten temat na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury. Z innych tematów, które zostały poruszone przez państwa posłów, szczególnie w zakresie BRD - drodzy państwo, jestem w stanie przekazać statystyki, które mamy, jeżeli chodzi o pierwsze 5 miesięcy roku 2019, dotyczące liczby wypadków oraz zdarzeń na polskich drogach. Generalny spadek to spadek o ok. 20%. Spadek liczby wypadków - minus 25%. Spadek liczby kolizji - minus 23%. Cały czas inwestujemy w infrastrukturę, nie tylko w sieci dróg szybkiego ruchu. To blisko 500 tytułów inwestycyjnych na sieci już istniejącej: chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji pani minister Wanda Buk. Bardzo proszę, pani minister. Wysoka Izbo! Wynotowałam sobie po kolei pytania, które padały, dotyczące cyfryzacji.

Dalszych zmian w tym zakresie nie przewidujemy.

Szanowni państwo, muszę państwu powiedzieć, że jesteśmy ewenementem w Europie: mamy numer rejestracyjny zarówno na tablicach rejestracyjnych, jak i na naklejce. To jest wydatek dla obywatela zupełnie zbędny.

Oczywiście będą stopniowo dodawane kolejne funkcjonalności.

Dziękuję bardzo, pani minister. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Pani Minister! Wyjaśniam, że nie chodziło o przypadki dotyczące pojazdów, które zostały wyrejestrowane i są oznaczone w bazie centralnej ewidencji pojazdów jako archiwalne, bo wszyscy wiemy, że tak jest. Ja pytałem o sytuację, w której pojazdy nie istnieją, nie jest płacone za nie obowiązkowe ubezpieczenie, natomiast nie zostały wyrejestrowane i w bazie CEPiK istnieją jako funkcjonujące.

Jeżeli państwo nie są gotowi, to poproszę o odpowiedź na piśmie, może nawet lepiej, gdyby to było na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Na piśmie.

Dobrze, bardzo proszę. Szanowna Pani Minister! Pragnę panią zapewnić, że nie pytałem pani o kwestię dotyczącą naklejek i nie jestem zwolennikiem dodatkowego obciążania obywateli naszego kraju jakimikolwiek opłatami wtedy, kiedy tych opłat być nie powinno. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 388, do Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Ogłaszam przerwę do godz. 17.30. Dziękuję.

Wznawiam obrady. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym oraz poselskim projekcie ustawy o instrumencie wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych w zakresie realizacji planów wypoczynkowych w latach 2020–2022 w związku z pandemią COVID-19, druk nr 429. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Marszałek Sejmu proponuje, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Panie Ministrze! Szanowni Posłowie! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o instrumencie wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych w zakresie realizacji planów wypoczynkowych w latach 2020–2022 w związku z pandemią COVID-19, druk nr 422, oraz o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, druk nr 423. Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 429. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 18 czerwca 2020 r. projekt ustawy z druku nr 422 do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przeprowadziła w dniu dzisiejszym pierwsze czytanie. Oba projekty były poddane pierwszemu czytaniu, przy czym projekt z druku nr 423 był drukiem podstawowym. Szanowni Państwo! Można powiedzieć, że poprawki są związane z wprowadzeniem bonu turystycznego, który ma na celu dalsze wsparcie branży turystycznej ponoszącej bardzo duże ujemne efekty zatrzymania ruchu turystycznego w Polsce, oraz z tą przesłanką, która towarzyszyła i Prawu i Sprawiedliwości, i panu prezydentowi przez poprzednie lata, które są już za nami, zdecydowanego wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci. W związku z tym te dwa cele w ustawie o bonie turystycznym bardzo mocno się spinają, wiążą i oba te cele będą osiągnięte. Pamiętajcie państwo, ponieważ ja jestem człowiekiem z edukacji, jak wiele czasu poświęcaliśmy w komisjach, żeby dzieci jeździły na wycieczki szkolne, ponieważ nie ma w zasadzie takich środowisk, w których wszystkie dzieci stać na to, żeby pojechać na wycieczkę historyczną. Teraz jest ta szansa. Pięknie szkoły będą mogły razem z rodzicami te środki kierować również na cele edukacyjne.

Kolejne poprawki dotyczyły podniesienia wartości bonu, przeważnie dwukrotnie. Również nie uzyskały one poparcia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja przyjęła dwie poprawki.

Jest ich dziewięć. Wnoszę, aby Wysoki Sejm raczył uchwalić załączony projekt ustawy. Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pani poseł Urszula Rusecka. Bardzo proszę, pani poseł. Pani Marszałek! Pani Minister! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec przedstawionego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym z druku nr 423. Panie Prezydencie! Bardzo dziękujemy za polski bon turystyczny zapowiadany i dyskutowany już na początku kwietnia. To kolejny przykład wiarygodności i dotrzymywania słowa danego Polakom przez pana prezydenta.

Obok instrumentów zawartych w tarczy antykryzysowej i finansowej to kolejny program dedykowany tej branży. Należy podkreślić, że polski bon turystyczny po raz kolejny wychodzi naprzeciw potrzebom polskich rodzin, stanowiąc realne wsparcie w organizacji i finansowaniu wypoczynku ok. 6 mln dzieci, w tym 300 tys. dzieci z niepełnosprawnościami. To dobrze, że w projekcie zostały zawarte także zapisy pozwalające na wsparcie dla samorządów w prowadzeniu i finansowaniu przez nie inwestycji. Beneficjentami ustawy będą wszyscy przedsiębiorcy turystyczni, począwszy od gospodarstw agroturystycznych, na hotelach kończąc. Na uwagę zasługuje kwota 4 mld zł, które dotychczas zostały przekazane branży turystycznej w ramach wszystkich tarcz, co stanowiło realną pomoc dla ok. 15 tys. beneficjentów. Tylko dzięki ogromnemu wysiłkowi oraz dobrej współpracy rządu Zjednoczonej Prawicy i prezydenta Andrzeja Dudy udaje się Polskę bezpiecznie przeprowadzić przez światowy kryzys. Głównym czynnikiem decydującym o znacznym ograniczeniu strat gospodarczych związanych z wirusem była szybka reakcja polskiego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, na to, co zadziało się w świecie. Duży pakiet pomocowy uchronił polskie firmy od bankructw i poważnej utraty miejsc pracy. Przypomnę, że na dzień dzisiejszy bezrobotnych jest niecały 1 mln, natomiast jeszcze w 2015 r. bezrobotnych było prawie 2 mln. Szanowni Państwo! Prezydent Andrzej Duda wraz z rządem Zjednoczonej Prawicy poprzez przełomowe społeczne i solidarnościowe programy inwestuje w polskie rodziny, w polski biznes. Ta ustawa jest kolejnym takim programem, który będzie wspierał polskie rodziny. Bardzo dziękujemy jeszcze raz za tę ustawę i wierzymy w to, że będzie dobrze służyć i polskim rodzinom, i branży turystycznej, ale nie jest to jeszcze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o branżę turystyczną. Kolejne programy dla tej branży są już w przygotowaniu, bo wiemy, że ta branża jest jedną z tych branż, które najbardziej ucierpiały z powodu światowej epidemii. Klub Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie opiniuje powyższą ustawę. Szanowna pani marszałek, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość składam wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, druki nr 422, 423 i 429, bez odsyłania do komisji poprawek i wniosków zgłoszonych do tego projektu ustawy i o doręczenie ich posłom. Dziękuję, pani poseł. Dziękuję bardzo. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Ireneusz Raś. Wysoki Sejmie! Oczywiście nie zgadzam się z tym, że jest to przełomowy projekt, program. To jest program minimalny, dlatego moje środowisko polityczne mimo niepodjęcia w ogóle debaty nad naszym projektem, projektem powszechnym, jeżeli chodzi o kierowanie tego programu do polskiego biznesu turystycznego, jeżeli chodzi o Polaków, nie chciało dzielić, chciało uruchomić energię Polaków, żeby ona uratowała w perspektywie najbliższych miesięcy, najbliższych 2 lat, potencjał polskiej gospodarki turystycznej, polskich przedsiębiorstw turystycznych. Z taką skalą mamy do czynienia. Dziś to, co państwo proponujecie, po analizie.

W niektórych wypowiedziach jej współpracowników padały kwoty 9 mld zł.

Dziś mamy sytuację nadzwyczajną, czyli środków powinno być więcej.

To dość duża zgoda.

Być może, jeśli będziemy tam dokładać perspektywy, to ta branża z tego mechanizmu, który jeszcze, mam nadzieję, ulegnie zmianie po spokojnej debacie, a nie w piku kampanii wyborczej, w Senacie.

Dziękuję, panie pośle. Stanowisko klubu parlamentarnego Lewica przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Dariusz Wieczorek. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rzeczywiście przebieg tej dyskusji w komisji wskazuje na jedną rzecz. Ktoś zostawił długopis, pewnie pan poseł. No to tutaj zostawiam. A, może tak. Rzeczywiście tak się dzieje w naszym kraju w ostatnim czasie, że właściwie rząd nie jest potrzebny. Wystarczy nam prezydent, bo prezydent wszystko inicjuje: i dodatek solidarnościowy, i bon turystyczny. Oczywiście prawda jest taka, Lewica mówi to jasno i wprost, że lepiej jest coś mieć, niż nie mieć nic. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale żeby była jasność - pani poseł sprawozdawca już to powiedziała - te kwoty, które tutaj są podane, 4 mld zł, to jest kropla w morzu potrzeb, jeżeli chodzi o ratowanie branży turystycznej.

W turystyce jeżeli w marcu, w kwietniu, w maju nie sprzedano miejsca noclegowego, to to już nie wróci. Padały różne kwoty dotyczące tych wpływów.

W związku z czym w tym zakresie rzeczywiście byłaby potrzeba, żeby tę pomoc ewidentnie zwiększyć.

Pytanie jest takie. Znowu mamy kolejne obciążenie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sensie dodatkowej pracy, mamy dodatkowe obciążenie dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Enigmatycznie napisano, że oczywiście z tego funduszu te dodatkowe koszty będą pokrywane, ale znowu musimy zwrócić uwagę na to, że te instytucje będą miały dodatkowe zadania, podobnie jak pewne zadania będą miały samorządy. W związku z tym to najlepiej świadczy, w jakiej procedurze jest ten projekt przygotowywany. Ani z branżą turystyczną, ani z samorządami to nie było po prostu konsultowane. I to jest też zarzut do państwa, że robicie to szybko, w tym szale wyborczym, i tu oczywiście można w tym zakresie popełnić dużo więcej błędów, niż rozmawiając i dyskutując z samymi zainteresowanymi. Oczywiście pojawiła się też zmiana... bo to już jest w tych wszystkich ustawach COVID-owych, to jest właśnie bardzo ciekawa rzecz, że one zmieniają na ogół 40 innych ustaw. I jest propozycja, poprawka, o której pani poseł sprawozdawca mówiła - pojawia się wsparcie na zadania inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego. Super, to jest dobre rozwiązanie, tylko znowu: jeżeli decyzje w tej sprawie ma podejmować rząd i ma w tej sprawie podejmować uchwałę, to chcielibyśmy wiedzieć, jaki jest planowany zakres tej pomocy na te zadania inwestycyjne dla samorządów, żeby znowu nie było to w jakiś sposób nieuczciwy wykorzystywane. Kończąc - były pewne zastrzeżenia Biura Legislacyjnego do naszych poprawek, one znalazły się wśród poprawek mniejszości. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Państwo Ministrowie! Szanowni Panowie! Rozmawialiśmy dzisiaj w komisji o propozycji pana prezydenta. Ubolewam, jak już mój przedmówca powiedział, że nie miała takiej okazji, szansy komisja kierunkowa - komisja turystyki. A turystyka mówi dzisiaj, że potrzebuje wakacji leasingowych, kredytowych na kolejny okres.

Branża turystyczna, szanowni państwo, dzisiaj dzięki bonowi turystycznemu nie odbije się.

My dzisiaj obserwujemy, jak wielkie trudności napotyka właśnie ten obszar. To, że zostały uruchomione niektóre działania, nie znaczy, że z dnia na dzień można było uzyskać efekty. Pani premier mówiła dzisiaj, jak dużo PKB jest właśnie z tej dziedziny, ile osób pracuje w turystyce. To wsparcie, które zostało wygenerowane, pani premier, musi trwać dłużej. Są branże, które po prostu nie podźwigną się, i to jest bardzo potrzebne. Pomysł pana prezydenta, zgodzę się tutaj z moimi przedmówcami, jest bardzo mocno wyborczy.

Później jest troszeczkę inaczej. Ten projekt, szanowni państwo, powtórzę to po raz kolejny, dzieli Polaków. On nie powinien dzielić, on powinien łączyć Polaków. Dlatego my jako Klub Parlamentarny Koalicja Polska złożymy kolejne poprawki. Choćby związaną z tym, szanowni państwo, że przypisaliście te pieniądze tylko i wyłącznie do dzieci, a czasami bywa tak, że w niektórych hotelach czy w przypadku usług gastronomicznych te dzieci są zwolnione z pewnych opłat. Ale już nie będzie obowiązywał bon.

I może, szanowni państwo, byłoby lepiej, gdyby pan prezydent nie pojechał do tych Stanów Zjednoczonych, bo to nas znowu będzie kosztowało, Polaków, kilka miliardów złotych - kilka miliardów złotych. Może lepiej by było zgodzić się z tymi, którzy mówią, że prezydent powinien w Polsce zostać, i zająć się wreszcie tymi rzeczami, które Polaków interesują i które Polakom przeszkadzają. Mam nadzieję, że będziemy mogli dalej dyskutować.

Fundusz płynności dla turystyki - to jest właśnie to rozwiązanie. W imienia Koła Poselskiego Konfederacja głos zabierze pan poseł Jakub Kulesza. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wiele się ostatnio mówi o niszczeniu polskiej rodziny i trzeba to powiedzieć wprost: to państwo niszczą polską rodzinę, bo to państwo niszczą polską gospodarkę podatkami, inflacją, zadłużaniem przyszłych pokoleń.

No i wybory prezydenckie 10 maja - 10 dni wcześniej miała być wypłacona kolejna trzynasta emerytura, ale że wybory się przesunęły, to musieli państwo wymyślić następne rozdawnictwo, no i jest 500+ w postaci bonu turystycznego.

Ja wiem, kto jest winny - Platforma Obywatelska, naprawdę. Popatrzcie, trzy ostatnie programy: trzynasta emerytura, 500+ na każde dziecko i bon turystyczny. Kto to wymyślił i obiecał? Skoro łżekonserwatyści i łżeliberałowie realizują zgniły program socjaldemokracji, to po co nam Lewica? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.

Życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy oferują usługi i eventy turystyczne, ale ten projekt, była o tym mowa, to przekupstwo przedwyborcze i na dodatek selekcjonujące Polaków, dzielące ich, jak to u socjalistów, na gorszych i lepszych.

Ten projekt, którego posłowie nie dostali wcześniej, tłumacząc z polskiego na nasze, to jest taka tarcza 5+ turbo dla rządu.

Dopiero po chwili dotarło do mnie, że to jest poprawka helikopterowa, że to jest właśnie ten helikopter dla pani premier, żeby mogła latać nad Polską i rozsypywać dywanowe pieniądze. precyzuje i wyraźnie artykułuje.

Regulaminowo złożyłem tę poprawkę przewodniczącej komisji, która nieregulaminowo i bezprawnie nie poddała tej poprawki pod głosowanie. Procedujcie, procedujcie, głosujcie.

Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytań. Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Przemysław Koperski, klub Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Premierze!

To dzisiaj ok. 170 tys. zł. I pytanie: Czy jesteście na to przygotowani? Dzisiaj tyle wynosi maksymalna kara administracyjna dla mieszkańców województwa śląskiego, którzy zostali przyłapani w Republice Czeskiej, również ci podróżujący wakacyjnym tranzytem do Austrii czy Chorwacji. I to jest nienormalna sytuacja. Panie Premierze Morawiecki! Chcę się dowiedzieć, czy w końcu pan wykona telefon do Andrzeja Babisa. Chciałbym też zapytać ministra zdrowia Szumowskiego, czy.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

To są takie miejscowości, gdzie jest wielu małych, średnich przedsiębiorców turystycznych. I oczywiście, jeśli popatrzymy na propozycję pana prezydenta, lepiej mieć coś niż nie mieć nic, chociaż muszę powiedzieć, że przedsiębiorcy sami sobie co najmniej w połowie zapłacą za to wsparcie, bo przecież płacą podatki: VAT, podatek dochodowy. Natomiast myślę, że dzisiaj trzeba zadać zupełnie inne pytanie, bo w województwie śląskim, o czym mówił mój przedmówca, mamy dzisiaj potężny kłopot z relacją z naszymi przyjaciółmi Czechami.

Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rozmawiamy o bonie turystycznym, ale chciałbym Wysokiej Izbie przypomnieć, że w Polsce żyją również emeryci i renciści. Mamy, szanowni państwo, najnowsze dane. Po marcowej waloryzacji okazało się, że w Polsce 333 tys. emerytów nie otrzymuje emerytury minimalnej. Szanowni Państwo! Panie Ministrze! Jak to się stało, że w planach wypoczynkowych Polaków zapomnieliście o tej grupie społecznej? Dlaczego ją wykluczacie? Dlaczego emeryci, którzy są również najbardziej skazani na skrajną biedę, na skrajne ubóstwo, które rośnie w tej grupie wiekowej, w tej chwili wykluczani są z możliwości po okresie zagrożenia epidemicznego, stanie epidemii, tak naprawdę są uwięzieni w swoich mieszkaniach? Dlaczego wykluczacie emerytów? Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bon 500+, bon turystyczny, mimo że jest wsparciem potrzebnym dla branży turystycznej, jest również potwierdzeniem prowadzonej od lat przez rząd Prawa i Sprawiedliwości polityki wykluczenia. Gdzie zatem ci wszyscy, którzy dziś płacą podatki? Gdzie osoby nieposiadające dzieci, gdzie emeryci i renciści, gdzie młodzi ludzie płacący podatki, gdzie studenci?

Dlaczego wyłączacie z tego projektu kolejne grupy społeczne?

Bardzo proszę.

Mamy do czynienia tak naprawdę z jednorazową waloryzacją tracącego na wartości wskutek ciągłego wzrostu cen świadczenia 500+. W uzasadnieniu czytamy także, że przyznanie rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych dodatkowego świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł jest formą realnego, efektywnego, instytucjonalnego wsparcia. Szkoda tylko, że o niepełnosprawnych przypomina się rządzącym wyłącznie przed wyborami. Tak niestety jest. Potrzebny jest plan odbudowy wypracowany wspólnie przez branżę i przez rząd. Gdzie konsultacje społeczne? Bardzo proszę. Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! W ostatnich tygodniach głośno było na temat inicjatywy pani wicepremier Jadwigi Emilewicz wprowadzenia bonu turystycznego w wysokości 1 tys. zł. Jak się wkrótce okazało, rząd z pomysłu się wycofał. Dlatego ze zdziwieniem przyjąłem wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, zresztą na wiecu wyborczym, że każda rodzina jeszcze przed wakacjami otrzyma bon turystyczny na wzór programu 500+ na każde dziecko. Pomysł ten o tyle zaskakuje, że to już drugi projekt po dodatku solidarnościowym, który prezydent chce zrealizować tuż przed wyborami. W związku z powyższym dlaczego rząd wycofał się ze swojego pierwotnego pomysłu? Czy odpowiedź jest po prostu taka, że rząd zamierza po raz drugi po przyjęciu dodatku solidarnościowego wesprzeć kolejny raz pana prezydenta w kampanii wyborczej? Dlaczego nie wzięto pod uwagę propozycji Koalicji Obywatelskiej, która obejmowała nie tylko dzieci, ale m.in. osoby (Dzwonek) starsze? Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ale, proszę państwa, Polska starzeje się, za 2 dekady będziemy drugą Florydą, miejscem, gdzie ogromną większość stanowią emeryci. Tak więc kiedy program wspierający zwiększenie dzietności w Polsce?

Tak że zwracam się do klubu Koalicji Obywatelskiej, żeby wpłynął na swoich radnych i uchwalił wsparcie dla osób mniej zamożnych w województwie podlaskim, w stolicy tego województwa. Bardzo proszę. Pani marszałek, czy możemy jeszcze jedno. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Gdańska Organizacja Turystyczna i Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna przeprowadziły badania, których celem była analiza skutków epidemii dla firm branży turystycznej województwa pomorskiego, tego województwa, którego jestem posłem. W badaniu udział wzięło 250 firm branży turystycznej. Większość, 63% firm, wskazała, że niezbędna jest pomoc finansowa zarówno ze strony rządu, jak i władz samorządowych. Postulaty w tym zakresie najczęściej dotyczyły zwolnień, obniżek lub rozłożenia w czasie płatności. Podatki lokalne - o tym wspomniało 38% respondentów, składki ZUS - 18, wsparcie w utrzymaniu pracowników - 12, czynsze - 10. Bon turystyczny w wysokości 500 zł jest dobrym zabiegiem przedwyborczym, jednak nie odpowiada na rzeczywiste potrzeby branży turystycznej i nie jest także wystarczającą, realną pomocą dla rodzin. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Zapewne jak i miliony Polek i Polaków znacie mem, na którym widnieje pies pijący sok z kartonu, na którym jest napis: sok dla kretynów. Opis tego zdjęcia: kiedy jesteś bezdzietnym, pracującym i niekaranym obywatelem powyżej 26. roku życia i wierzyłeś, że rząd ci da choć jedną rzecz, czyli ten bon na wakacje. Pytanie jest proste: Co wy na to?

Gdzie są emeryci i gdzie są pozostałe osoby, które również zasługują na te pieniądze, które wcześniej wypracowały? Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Niska zawartość mięsa w tej kiełbasie wyborczej, same skórki, ścinki i chrząstki, na grilla się nie nadaje. Jeszcze przed pandemią 40% dzieci nie korzystało z usług przedsiębiorstw turystycznych. Rodzin tych dzieci pomimo bonu nadal nie będzie stać na wysłanie dzieci na wypoczynek. Nie możecie się doliczyć, ile dzieci nie mogło korzystać ze zdalnego nauczania z braku komputera i Internetu, a to będą te same dzieci, których bony nie przejdą aktywacji w PUE ZUS. Z usług administracji publicznej za pomocą Internetu korzysta jedynie 40% obywateli, a to jeszcze gorzej wróży. No i zapomnieliście o emerytach. Zapomnieliście o emerytach, bo za dużo by was to kosztowało. Zapomnieliście także o instytucjach kultury, których wpływy własne w okresie pierwszych dwóch miesięcy pandemii wyniosły zero, a teraz nie ma przecież grup zorganizowanych, więc te wpływy są nadal mizerne. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To jest następna ustawa socjalna, taka jak 500+, trzynasta emerytura, czternasta emerytura. Do wszystkich tych z branży turystycznej teraz mówię: Nie myślcie, że pan prezydent pochylił się nad waszymi problemami. Nie, nie pochylił się, tak po prostu wyszło. Koronawirus złapał nas w okresie przedwakacyjnym, a więc dostaliśmy bon wakacyjny. Gdyby koronawirus złapał nas w okresie jesiennym, dostalibyśmy bon na węgiel. Tak to wygląda. Panie ministrze spraw wewnętrznych i administracji, do pana się zwracam. Tworzyć trzeba prawo dobrze. Pytam, dlaczego zapomniał pan o granicy wewnętrznej morskiej.

Proszę wreszcie, żebyście. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mamy kolejną ustawę. trzeba kupić głosy i obiecuje się najpierw 1 tys., później 500, 1 tys. dla wszystkich, 500 dla wszystkich. Okazuje się, że 500 dla wybranych. I dobrze, niech te dzieci pojadą, odpoczną. Ale co dalej? Szanowni państwo, branża turystyczna była wyłączona przez 3 miesiące zupełnie z funkcjonowania. Takie gminy np. jak Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Karpacz, Podgórzyn, do których nikt nie przyjeżdżał. Niestety nie miały jakichkolwiek przychodów, ponieważ przedsiębiorcy nie płacili CIT-u ani PIT-u, podatek od nieruchomości nie wpływał, bo ludzie nie mieli z czego zapłacić. Jak pomożemy tym mieszkańcom?

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Chciałbym wierzyć w to, że propozycja tej ustawy nie jest tylko i wyłącznie przedwyborczym trikiem. Kiedy pan prezydent podpisywał ustawę przekazującą 2 mld zł na TVP, obiecywał stworzenie funduszu zdrowotnego. Gdzie jest ten fundusz? Prezydent obiecywał podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Gdzie jest ta kwota? Nie ma. Prezydent obiecywał 100 tys. mieszkań dla młodych. Gdzie są te mieszkania? Nie ma. Prezydent obiecywał, że będziemy potęgą w budowie statków.

Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przypomnę, że 10 dni temu klub Koalicji Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt ustawy gwarantującej 500 zł na wyjazd turystyczny dla każdej Polki i każdego Polaka. Pan prezydent wczoraj złożył swój projekt ustawy gwarantującej 500 zł, ale tylko na dziecko. Pytam: Co z osobami, które nie mają dzieci? Dlaczego pan prezydent Duda o tych osobach zapomina? Dlaczego uważa, że pomoc tym osobom się nie należy?

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Pytanie, czy będzie na to stać biedne polskie rodziny. Ale zastanówmy się nad czymś jeszcze innym. Tu padnie pytanie: Co zrobić z rodzinami, które są wykluczone informatycznie? Jak one złożą wniosek o ten bon? Ile tych dzieci nie pojedzie? Te statystki są ogólnodostępne.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Premier! Chciałbym prosić panią premier o objaśnienie Wysokiej Izbie art. 43, który jako wrzutkę na zakończenie pracy nad projektem prezydenckim zgłoszono w trybie poselskim. Przedstawiciele Biura Legislacyjnego mówili o wadliwości tej procedury, o podejrzeniu o niekonstytucyjność, ale sprawa, której dotyczy ta poprawka, jest ważna. Chodzi o możliwość udzielania wsparcia na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządowych. Pytamy w takim układzie: Jakie zadania? Jaka kwota? Kiedy ten program będzie uruchomiony? Czy pani minister jest tak bardzo zapracowana, że nie była w stanie przygotować projektu rządowego w tak ważnej sprawie?

Bardzo proszę. Wysoka Izbo!

Dziś podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny prezydencki minister mówił, że bon turystyczny wesprze rodziny, ale przecież rodzina to nie tylko rodzina z dziećmi. To także rodzice, których dzieci są już dorosłe.

Co z tymi, którzy wychowali dzieci i ciężko pracują? Co z emerytami? Co ze studentami? Co z wszystkimi, którzy pracują, a nie posiadają dzieci? Im według waszego projektu bon turystyczny się nie należy.

Bardzo proszę. Nie ma. Bardzo proszę. Wysoka Izbo!

Dlaczego, panie prezydencie, nie pamiętał pan o emerytach i rencistach? Dlaczego nie pamiętał pan o tej grupie? Nasze Rodos - mówią - to nie jest Rodos poza granicami kraju, to są rodzinne ogrody działkowe i tylko to. Mam też jedno szczegółowe pytanie, mianowicie pytanie takie: Czy bon dla dzieci niepełnosprawnych będzie mógł być połączony z dotacją ze środków PFRON-u jako uzupełnienie wkładu własnego? To jest bardzo ważne. Ja dziwię się temu procedowaniu, które tutaj następuje, że nie zostało to przekazane do komisji turystyki. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! Pierwsze pytanie jest następujące. Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje kolejne zadanie. My stajemy, ja staję po stronie pracowników ZUS-u, którzy są naprawdę w tej chwili mocno obciążeni w wyniku tych ustaw, które zostały przyjęte, jeżeli chodzi o ustawy COVID-owe.

Rzeczywiście art. 43 mówi tak, że Rada Ministrów może określić, w drodze uchwały, zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zakres, sposób i termin przedstawiania tejże informacji.

Bardzo proszę. Pani Minister! Drugi miesiąc z rzędu spadają realne wynagrodzenia Polek i Polaków. Rynek pracy skurczył się o 270 tys. etatów. Wskaźnik dobrobytu Polek i Polaków zanotował gigantyczny spadek i jest już teraz niższy niż w 2009 r., a na pewno dołek jeszcze przed nami. Tymczasem pani minister cały czas jest w dobrym nastroju, chociaż zajmuje się pomocą doraźną zamiast systemową. Z drugiej strony wydaje się, że idzie druga fala epidemii, bo zamrożenie gospodarki na 2 miesiące, w tym także turystyki, problem tylko oddaliło. Liczba chorych i zgonów ponownie rośnie i średnia jest zapewne większa niż w maju, dzienna, w związku z czym chciałabym zapytać, dlaczego mogliśmy pojechać na weekend czerwcowy, pani minister, a nie mogliśmy pojechać na weekend majowy, skoro dzisiaj wzrost zachorowań jest większy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Bardzo serdecznie dziękuję, pani marszałek. Pani Premier! Te 500 zł, ten bon to dobry pomysł. Dobrze, że rząd zdecydował się na to, żeby poprzeć projekt prezydenta. o którym pracownicy, pracodawcy, ludzie, którzy z niego skorzystają, usłyszeli. Mam konkretne pytanie do pani premier, bo pani premier ma dobre serce i czasami pomaga, rzeczywiście chce. Czy da się, żebyśmy te 500 zł np. spróbowali obiecać na przyszły rok?

Ważne, żeby Polacy mogli na wakacje wyjeżdżać i wyjeżdżali. Pani premier - do pani, ale i do pana ministra Muchy. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. O głos poprosił zastępca szefa Kancelarii Prezydenta minister Paweł Mucha. Zapraszam serdecznie, panie ministrze. Szanowna Pani Premier! Wysoka Izbo! Tak, prezydent realizuje swoje obietnice, prezydent realizuje swój program. Tak, prezydent wykonuje swoją misję, swój urząd. Także wtedy, kiedy są potrzeby szczególne dotyczące kwestii związanych z walką z koronawirusem, skutkami społecznymi, ekonomicznymi i gospodarczymi, nie tylko zdrowotnymi, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podejmuje te wyzwania. Mamy sytuację specjalną. Mamy sytuację związaną z walką z pandemią światową, która dotknęła w szczególnym stopniu polskich przedsiębiorców, a wśród polskich przedsiębiorców - w szczególności branżę turystyczną. Wiemy, że to wsparcie dzisiaj dla branży turystycznej jest potrzebne. Stąd prezydent niezwłocznie podjął działania i skutkiem tych działań, podejmowanych w konsultacji z Ministerstwem Rozwoju, jest zaprezentowana państwu ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. To są rozwiązania dzisiaj oczekiwane przez polskich przedsiębiorców, ale to są też rozwiązania, wbrew temu, co tutaj mówiono, konsultowane ze środowiskiem polskich przedsiębiorców. Te prace, które były prowadzone, to są konsultacje, które były prowadzone bezpośrednio przez panią premier Jadwigę Emilewicz też, ale to są konsultacje, które prowadziła i Kancelaria Prezydenta bardzo szeroko. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, bezpośrednio współpracując czy to z Narodową Radą Rozwoju, czy z Radą ds. Przedsiębiorczości, czy z ekspertami, ale także spotykając się z Polakami w całej Polsce, w tym także z przedsiębiorcami turystycznymi, te założenia projektu konsultował na bieżąco. Efektem tej dyskusji jest przedłożona ustawa. To wsparcie ma podwójne umocowanie, bo z jednej strony to jest wsparcie, tak jak mówimy, dla przedsiębiorców, z drugiej strony, absolutnie macie państwo rację, to jest wsparcie dla polskiej rodziny. Jeżeli dzisiaj analizujemy treść Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i patrzymy na treść art. 18, który stanowi o szczególnym także wsparciu, ochronie rodziny, jeżeli patrzymy na przepis art. 68, gdzie jest mowa także o prawie do zdrowia, art. 69, który stanowi o wsparciu dla niepełnosprawnych, art. 71, który stanowi o priorytecie dla wsparcia dla rodziny, to te przepisy i te uwarunkowania konstytucyjne także są w tym projekcie odwzorowane.

Dla milionów polskich rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci, to jest więcej niż realizacja zapowiedzi, która się pojawiała w przestrzeni publicznej wcześniej, bo była mowa o 1 tys. zł na rodzinę. Natomiast wtedy kiedy była mowa o 1 tys. zł na rodzinę, była także mowa o uwzględnieniu w ramach finansowania tego programu współfinansowania ze strony pracodawców. Pojawiały się jednak takie głosy, które ostatecznie zostały wzięte w tym projekcie pod uwagę, że dzisiaj z uwagi na trudną sytuację, jeżeli chodzi o polskich przedsiębiorców, nie jest możliwe takie współfinansowanie.

Impreza turystyczna, usługi hotelarskie - to są pojęcia, które także zostały w tej ustawie zdefiniowane. Jeżeli chodzi o imprezę turystyczną, zdefiniowano ją bardzo szeroko: to będą turnusy rehabilitacyjne, to mogą być także wyjazdy, które są organizowane właśnie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci.

ZUS jest do tego przygotowany, żeby obsłużyć każdego potencjalnego beneficjenta takiego programu, czyli rodziców czy opiekunów prawnych tych dzieci. Uruchomiona zostanie także specjalna infolinia, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informację. Planujemy także szeroką akcję informacyjną.

Jeżeli chodzi o wsparcie dla Pomorza Zachodniego, to zwłaszcza takie powiaty jak: Świnoujście, kołobrzeski, kamieński, gryficki będą korzystać ze środków, które są przewidziane w tym programie.

Nam zależy na zrównoważonym rozwoju całej Polski, zależy nam na tym, żeby ludzie z mniejszych miejscowości, ze wsi, z miast mieli takie same, równe szanse i żeby Polska rozwijała się równomiernie. Ten program także, wbrew temu, co państwo mówicie, jest powszechny. On nikogo nie wyklucza. A naprawdę trzeba być ogromnie złej woli, żeby zapominać o wsparciu, które pan prezydent przewiduje dla emerytów. I tutaj można wymieniać takie programy jak: trzynasta emerytura, bezpłatne leki dla seniorów. Zapowiadam tę inicjatywę, o której pan prezydent też mówił, czyli Centrum Zdrowia 75+. Dzisiaj dochód przeciętnej rodziny, dochód rozporządzalny polskiej rodziny to jest absolutny priorytet, jeżeli chodzi o prezydenturę pana prezydenta Andrzeja Dudy, i my to wspólnie z polskim rządem realizujemy. Wzrosła stawka godzinowa, jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne, rośnie minimalne wynagrodzenie, rosną dochody, które są do dyspozycji polskiej rodziny. To jest ta szczególna troska pana prezydenta, który o to zabiega. Taki był jego program, który ogłaszał w 2015 r., i ten program konsekwentnie jest przez niego realizowany. 6 mln polskich dzieci skorzysta z tych rozwiązań, o których rozmawiamy, 300 tys. dzieci niepełnosprawnych. To 4 mld zł, które będą służyć właśnie przedsiębiorcom, którzy są aktywni w branży turystycznej. Tak jak powiedziałem, zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Polska Organizacja Turystyczna są gotowe do realizacji tej ustawy, która we współpracy z tymi podmiotami była przygotowana. Wbrew temu, co państwo mówicie, beneficjentami tego programu, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, w 85% - takie są szacunki - będą mikro- i mali przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, tę ustawę trzeba przyjąć, bo to są dobre rozwiązania. Szanowni państwo, takim bardzo wstrzemięźliwym, bym powiedział, głosem ujmę to tak: kwestie związane z zasadami, trybem udostępniania, realizacji czeku zostały odesłane do regulacji w drodze rozporządzenia. Ta delegacja miała charakter blankietowy, nie zawierała żadnych wytycznych co do sposobu regulowania tej kwestii. To była kiełbasa wyborcza, tylko przygotowana nieprofesjonalnie, na zasadzie blankietowego hasła bez żadnych analiz. Przecież jeżeli spojrzymy na te 6 mld zł, o których państwo mówicie, że miało zapewnić powszechny udział w tym czeku, i spojrzycie państwo na 4 mld zł, które zakładane są w tym projekcie prezydenckim, i spojrzycie, że tutaj jest tyle beneficjentów, ile wskazuje na to ustawa, 6 mln polskich dzieci, to ani rachunek ekonomiczny, ani żadna ocena skutków regulacji, ani żadne przepisy. Padały tu głosy, także posłów Lewicy, dotyczące obaw związanych z formułą elektroniczną, a państwo sami zakładaliście aplikację w tym zakresie. To jest tak, że te rozwiązania prawne, jeżeli zostaną przyjęte, a liczę na to, że zostaną przyjęte na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu.

O głos poprosiła również wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju pani premier Jadwiga Emilewicz. Bardzo proszę. Panie i Panowie Posłowie! Panie i Panowie Ministrowie! Przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim posłom za dzisiejszą wytężoną pracę nad tym projektem. Tak, zdajemy sobie sprawę, że pracujemy ponownie w tempie ekspresowym, ale takiego tempa dzisiaj wymaga od nas rynek, takiego tempa dziś wymaga od nas gospodarka. Również cieszę się, że zarzuty, które nam państwo tutaj postawili, są zarzutami o to, że realizujemy nasze obietnice. Taki jest znak szczególny obozu Zjednoczonej Prawicy, tak właśnie realizujemy programy, które deklarujemy.

Z taką konsekwencją realizujemy nasze programy. Powściągliwość i praca. Odnosząc się do wątpliwości i pytań, które tutaj padły, jak również dziękując i przyznając, że rzeczywiście Wysoka Izba w zgodzie przyjęła w pierwszej tarczy rozwiązanie dla branży turystycznej, które pozwoliło jej odsunąć w czasie spłatę należności za niewykonane usługi turystyczne, mamy nadzieję, że i tym razem w zgodzie przyjmiemy tę propozycję legislacyjną. Mówimy o tym, czy środki, które proponujemy, są dla branży wystarczające. Myślę, że możemy sobie powiedzieć jasno i otwarcie, że środki z tarczy, wszelkie środki pomocowe, które proponujemy, dzięki którym staramy się uratować możliwie jak najwięcej firm, zapewne nie trafią, nie będą wystarczające ani kompletne. Dlatego to nie jest nasze ostatnie słowo w zakresie branży turystycznej. Ten program przyczyni się do przetransferowania do branży 4 mld, niemal 4 mld zł, ale do niego należy dodać jeszcze 4 mld z tarczy finansowej, które już dzisiaj otrzymało ponad 15 tys. firm z branży turystycznej. Odpowiadając zatem na pytanie, dlaczego nie ma funduszu płynnościowego - to jest właśnie fundusz płynnościowy. Umarzalne pożyczki, umarzalne do wysokości 80%, w 3 dni dostępne na kontach przedsiębiorców - to jest realna pomoc, która od 29 kwietnia płynie do przedsiębiorców, w tym także do branży turystycznej. Ja zacytuję dziś tylko panią prof. Hannę Zawistowską ze Szkoły Głównej Handlowej, która powiedziała jasno: Najważniejsze w tym projekcie jest to, że środki trafiają bezpośrednio na konta i mają być adresowane bezpośrednio do branży turystycznej. Dzięki temu rodzice, na których wiele badań wskazuje, i tutaj dziękuję, bo jedna z pań posłanek o tym powiedziała, którzy w ogóle nie myślą nawet o tym, czy mogą dzieci wysłać na wakacje, będą mogli sfinansować obozy, obozy sportowe dla swoich dzieci, ponieważ to nie będzie wypłata na konto rodziców. To jest zatem nowoczesne rozwiązanie - odpowiadając na kolejne pytanie - które nie generuje nadmiernych środków kadrowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy w Polskiej Organizacji Turystycznej. Ono generuje wysiłek informatyczny i algorytmiczny, ponieważ to będzie kolejne rozwiązanie, które w sposób automatyczny będzie mogło być realizowane w punktach płatniczych. Zatem także za tym rozwiązaniem idzie kolejne unowocześnienie polskiego systemu administracji. Czy samorządy były konsultowane? Tak, rozmawialiśmy z samorządami. Od kilku tygodni jestem w stałym dialogu z organizacjami reprezentatywnymi, reprezentowanymi w komisji wspólnej rządu i samorządu. W trybie ekstraordynaryjnym, w trybie skróconym, ale tak, takie rozmowy prowadzimy. Robimy to nie, jak państwo mówią, w szale wyborczym, ale w stanie podgorączkowym pandemicznym, ponieważ my o tym rozwiązaniu mówiliśmy i analizowaliśmy to, a pan prezydent podjął się zadania przygotowania ustawy na początku kwietnia. ale mówmy o tym, kiedy projekt, który projekt jest gotowy do realizacji i kiedy będzie pierwsze świadczenie. I tak jak powiedział pan minister Mucha, jeśli Senat nie będzie zwlekał, to my jesteśmy gotowi organizacyjnie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polska Organizacja Turystyczna, aby w trzecim tygodniu lipca pierwsze płatności mogły być realizowane. Realizacja usługi na rzecz dzieci w hotelach. Oczywiście płacimy za hotel, czy jestem rodzicem z dzieckiem. Oczywiście za dziecko zwolnione z opłaty w hotelu rodzic będzie mógł zapłacić, ponieważ to nie jest przypisane do dziecka. Posiadanie dziecka jest kartą wstępu do świadczenia, natomiast świadczenie służy... to jest świadczenie rodzinne.

chyba państwo nie znają danych. Tak, jest wiele elementów, które się na to składają, także obniżona cena za baryłkę ropy, ale takie są dzisiaj dane. To są dzisiaj realne fakty, to jest ten moment, który upoważnia nas do tego, aby podejmować ambitne programy społeczne, aby podejmować ambitne programy gospodarcze, i dlatego to robimy. Właśnie może dlatego, że to nie jest kiełbasa wyborcza, tylko realny program pomocowy z jednej strony dla branży turystycznej, a z drugiej strony dla wsparcia rodzin. Przypomnijmy, ten bon trafi do ponad 6 mln dzieci, 6,4 mln dzieci to są beneficjenci tego programu.

Wspieramy w ten sposób głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, o których mówił pan minister Mucha, i mamy nadzieję, że za sprawą m.in. tego programu uda nam się utrzymać tętno polskiego sektora turystycznego. A mówimy, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Odpowiadając już na ostatnie pytanie, które zostało tutaj postawione, czy jest szansa na prolongatę. Myślę, że będziemy mogli, ponieważ my, kiedy zaczynaliśmy rozmawiać o instrumentach wsparcia polskiej branży turystycznej, myśleliśmy na początku tego roku, jeszcze przed stanem pandemii, mówiliśmy o pewnych trwałych rozwiązaniach, które są potrzebne. Robiliśmy analizę, jakiego rodzaju wsparcie dla branży turystycznej oferują inne państwa i w Europie, i poza nią. I mamy nadzieję, że jeżeli ten rok zakończymy z takimi perspektywami, o jakich dziś mówią eksperci międzynarodowi, że polska gospodarka będzie tą, która w najmniejszym stopniu ucierpi z powodu skutków pandemii ze względu na to, że zaoferowała szybką, skuteczną i celną pomoc, wówczas będziemy w stanie mówić o tym, że taki program będziemy mogli przedłużyć na kolejne lata, że on wpisze się w krajobraz wsparcia i wpisze się w rozwój branży turystycznej, ponieważ ona jest wizytówką i często otwiera bramy dla dużych, poważnych inwestorów. Tak rozumiemy naszą misję, tak rozumiemy nasze zadanie. Dzisiaj ono wymaga szybkich decyzji, i o takie szybkie decyzje dziś apelujemy i państwa prosimy. Tak jak państwu dziś rano wspomniałam, jesteśmy w stałym dialogu z branżą, rozmawiamy z przedstawicielami szeroko rozumianego sektora. Tak, wiemy, że dziś branża potrzebuje kredytów, że gwarancje de minimis z BGK do 80% są dla tej branży zbyt małe. Dlatego dziś pracujemy nad pakietem, który pozwoli gwarantować pożyczki w jeszcze nieco większym stopniu niż 80%. Mówiłam państwu także o wrześniu, który będzie trudnym okresem zwrotu za te usługi. I z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych także mamy już pewne założenia zmian. Tak jak powiedziałam: mniej mówimy, więcej pracujemy, przynosimy dobrze opracowane rozwiązania i liczymy na państwa współpracę w tym zakresie. Dziękuję bardzo, pani premier. Zamykam dyskusję. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Skoro mamy sprzeciw, do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań. Dziękuję.

Wznawiam obrady. Proszę państwa, ponieważ jesteśmy przed blokiem głosowań, przystąpimy do sprawdzenia kworum. Bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu stwierdzenia kworum. Bardzo proszę. Wiem, że nie działa, bo mój też nie działa.

Stwierdzam kworum. Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Uchwała Senatu to druk nr 426. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tej uchwały. Proponuję, na podstawie art. 54 ust. 8 regulaminu Sejmu, rozpatrzenie uchwały bez uprzedniego skierowania jej do komisji. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, druk nr 441. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 425. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Prezydium Sejmu, w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów, przedłożyło projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz oraz uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, druk nr 424. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego projektu. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz oraz uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (druk nr 424) Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz oraz uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. 14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie wyruszył transport polskich obywateli do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Wśród 728 pierwszych więźniów byli zarówno działacze polityczni, żołnierze kampanii wrześniowej, urzędnicy państwowi, nauczyciele, prawnicy, księża, jak i młodzież - harcerze, maturzyści i studenci. Data ich przyjazdu oznaczała początek funkcjonowania obozu zagłady w Auschwitz-Birkenau, który stał się symbolem niewyobrażalnego okrucieństwa i ludobójstwa. Droga, w którą wyruszyli więźniowie, dla większości z nich okazała się bezpowrotna - piekło obozu przeżyło niewielu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił w 2006 roku dzień 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Naszym obowiązkiem jest upamiętnianie wydarzeń, które miały miejsce na ziemiach okupowanych przez hitlerowskie Niemcy. Holokaust, zniewolenie i eksterminacja Polaków, Żydów, Romów oraz przedstawicieli wielu innych narodów są dla nas przestrogą i zobowiązaniem do działań, które sprawią, że ponowne zaistnienie takich zbrodni nie będzie możliwe. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć wszystkim ofiarom niemieckich nazistowskich obozów śmierci” Proponuję, żebyśmy przyjęli tę uchwałę przez aklamację. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz oraz uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (druk nr 426) Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. Senat proponuje zmianę odesłania do przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Głosowało 441 posłów. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

Sejm poprawkę odrzucił.

W 5. poprawce do art. 11 Senat proponuje w odesłaniu przytoczenie całego tytułu ustawy wraz z oznaczeniem rocznika.

Senat proponuje, aby wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosiła 1500 zł miesięcznie. Proponuję, aby Sejm wyraził zgodę na łączne głosowanie nad poprawkami od 6. do 9. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek od 6. do 9., zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym i senackim projektach ustaw o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 419-A. Proszę panią poseł Urszulę Rusecką o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Przypadło mi w udziale przedstawienie dodatkowego sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, druk nr 418, oraz o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, druk nr 283.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 419. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm będzie głosować w pierwszej kolejności. Nad tymi poprawkami będziemy głosować łącznie. Głosujemy. Kto się wstrzymał?

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 2. i 3., zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 419, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 417-A. Proszę pana posła Kazimierza Smolińskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Wysoka Izbo! Dodatkowe sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, druk nr 415. Sejm na posiedzeniu w dniu 19 czerwca skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 417 do komisji w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 417. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Sejm poprawki odrzucił. W 4. poprawce do art. 2 ustawy nowelizującej wnioskodawcy proponują nowe brzmienie przepisu przejściowego. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 417, wraz z przyjętą poprawką, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu oraz o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania bez odsyłania projektu do komisji. W pierwszej kolejności poddam pod głosowanie wniosek o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu uchwały zawartego w druku nr 421, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu uchwały zawartego w druku nr 421, zechce nacisnąć

Sejm wniosek przyjął. Przystępujemy zatem do drugiego czytania projektu uchwały. Pan poseł Braun. Proszę bardzo, panie pośle.

Bardzo proszę, panie pośle, 2 minuty.

Głosujmy sprzeciw. Kto jest za 2-minutowymi oświadczeniami w imieniu klubów i koła, proszę o naciśnięcie przycisku. Wiem, że nie działa. Działa. Kto jest za moją propozycją 2-minutowych oświadczeń? Kto jest przeciw?

Sejm propozycję przyjął. W związku z tym otwieram dyskusję, do której zgłosił się pan poseł Braun.

Szanowni Państwo! Wprowadziliście tutaj reżim, którego jeszcze w historii nowożytnej, tzn. postpeerelowskiej historii, tej Izby nie było. Za zmianami regulaminowymi, które wpisaliście tam z litery, poszły w praktyce rozwiązania nigdzie niezapisane, a uwłaczające powadze tej procedury, w której wszyscy uczestniczymy. Tego jeszcze nie było, żeby przed posłami zamykali i, reglamentując dostęp, otwierali drzwi członkowie, znakomitej zresztą, Straży Marszałkowskiej, po szereg żenujących sytuacji związanych z reglamentowaniem dostępu do tej mównicy, ale także reglamentowaniem czasu.

Nie przedłużajcie państwo tego stanu, nie przedłużajcie, nie kontynuujcie.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Wy to wiecie, więc ja wam nie będę mówił, będę bardziej mówił do obywateli, Polaków, którzy nas w tym momencie słuchają. Śpią tutaj za darmo w hotelu albo w mieszkaniu. Jedzą tutaj, w restauracji i w bufecie, za 1/3 ceny rynkowej, więc właściwie też można uznać, że jest to za darmo. Jedyne, co muszą posłowie zrobić, to przyjechać tutaj, do tej Izby, i tutaj siedzieć, w tych miejscach, gdzie mają się zebrać i gdzie mają głosować, gdzie mają decydować o tym, co będzie w państwie, gdzie mają zarządzać Polską. I Prawo i Sprawiedliwość właśnie dzisiaj mówi nam o tym, że im się tego nie chce robić, wolą robić to z domu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Do tych posłów, którzy siedzą w szlafroku na kanapie z tabletem w ręku: Ale ja wam powiem jedno: Do roboty. W pociąg, przyjechać tu, siedzieć.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość chciałbym poprzeć wniosek, projekt przedstawiony przez panią poseł w pierwotnym kształcie.

Uznaliśmy, że należy te przepisy wprowadzić na okres przejściowy, do końca czerwca.

I gdybyśmy tego przepisu nie wprowadzili, może dojść do paraliżu państwa, paraliżu Wysokiej Izby. Pamiętacie państwo, jak chcieliśmy zmienić regulamin, jaki był wówczas problem, że Wysoka Izba musiała się stawić - wszyscy musieli się stawić, większość - żeby przegłosować możliwość zdalnego głosowania. Jak wówczas przegłosujemy regulamin, żeby wrócić do zdalnego głosowania? Dlatego musimy zdecydować o tym, że przywracamy ten pierwotny kształt regulaminu Sejmu, że w sytuacji, w której obowiązuje stan wyjątkowy lub stan pandemii, pani marszałek może zdecydować o zdalnym głosowaniu lub też nie. I proszę wziąć pod uwagę właśnie kwestię bezpieczeństwa i państwa. Niektórzy z państwa nawet jeszcze ani razu nie byli na posiedzeniu Sejmu, są osobami starszymi, są osobami zagrożonymi. Dlaczego chcecie ich zmuszać do przyjazdu tutaj, a nie umożliwić im zdalne głosowanie? Proszę im to umożliwić dla ich własnego bezpieczeństwa. Pan poseł, który mówił o zagrożeniach związanych z komisjami tajnymi, że tu w sposób tajny. Przecież posiedzenia tajne się odbywają, panie pośle, różnego rodzaju, są komisje tajne. Tak że tu nie ma problemu, że Sejm nie obraduje w sposób tajny. W imieniu klubu parlamentarnego Lewica pan poseł. Proszę. Panie i Panowie Posłowie! Wstyd. Wstyd. Ja tu jestem na każdym posiedzeniu i żyję, panie pośle, i żyję. Wam Sejm przeszkadza. Wy z Sejmu chcecie zrobić przybudówkę rządu. Już wam to powiedziałam podczas pierwszego głosowania. A Sejm nie jest przybudówką rządu. Sejm ma was kontrolować. Sejm ma obradować na posiedzeniach. Wy się naprawdę, proszę państwa, brzydko bawicie, bo się bawicie konstytucją. Dzisiaj słyszałam od waszego prezydenta. Ale wy tę konstytucję depczecie i plujecie na nią każdego dnia tutaj, w tym Sejmie. I proszę nam nie opowiadać, że to jakby jest pandemia albo stan wyjątkowy. A kto decyduje, że jest pandemia albo stan wyjątkowy? Wy naprawdę. Zaczęło się nawet niewinnie: nocne głosowania, 30 sekund na pytania, przemówienia bez żadnego trybu. A jak się kończy? Wygaszacie Sejm. Chcecie się nas pozbyć, bo wam przeszkadzamy, bo się nas boicie. Bo się tutaj nas boicie. Panie marszałku, to dobrze, bo wolałabym pani marszałek tego nie powiedzieć. Po was to zamiast Sejmu zostaną te barierki i ta policja.

Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pani minister Emilewicz: Czy pani mnie słyszy? W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie Polaków [[Oklaski]] klub Lewica od samego początku stanu zagrożenia epidemicznego i późniejszego stanu epidemii wspierał wszystkie działania rządu zmierzające do ograniczenia skutków rozprzestrzeniania się COVID-19. Możliwość odbywania posiedzeń Sejmu, komisji i podkomisji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej niejednokrotnie przekraczała granice dobrego parlamentarnego obyczaju.

W takich warunkach nie da się zaplanować rzetelnej, uczciwej pracy w okręgach, nie da się uczciwie i odpowiedzialnie przygotować do obrad czy prac w komisjach. Apeluję do posłów i posłanek PiS-u, aby brali przykład z pana prezesa Kaczyńskiego, który na sali jest zawsze, natomiast tutaj zawsze jest wolna przestrzeń. Wiele zastrzeżeń mamy do pracy w komisjach. Prace w komisjach wyglądają bardzo źle: trzy, cztery osoby w 30-osobowych komisjach, reszta zdalnie, z tabletów, jedząc posiłek, może kosząc trawę w swoich posiadłościach. Lewica stanowczo opowiada się za przywróceniem obrad w Sejmie w trybie sprzed epidemii.

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 421, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysoka Izbo!

Co 3 miesiące premier miał składać informację.

Pan ma świadomość, że to nie jest wniosek formalny, prawda? Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druki nr 427 i 441) Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 441. Senat w swojej uchwale zaproponował do ustawy 126 poprawek.

Głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Przystępujemy do głosowania w związku ze sprzeciwem. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem przedstawionej przed chwilą propozycji dotyczącej sposobu głosowania nad poprawkami Senatu, zechce nacisnąć przycisk. jest przeciw?

Sejm propozycję przyjął.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Będzie wynik głosowania, to panu powtórzę.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 10. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 13. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 18. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem wymienionych poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Z poprawką tą łączy się poprawka 105. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 35. i 105., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawki Senatu bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 37. i 112., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawki Senatu bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 48. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Z poprawką tą łączy się poprawka 115. Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 60. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Jeszcze raz czytam. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 60. poprawki? się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. W 67. poprawce Senat proponuje skreślić pkt 6. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 67. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 76. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 84. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Z poprawką tą łączy się poprawka 120. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 89. i 120., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 94. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 97. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 98. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 109. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? To nie koniec głosowań, proszę państwa, więc proszę nie wychodzić.

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Powracamy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:

Poddam pod głosowanie wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez odsyłania do komisji. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm skierował projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy zawartego w druku nr 429, po doręczeniu zestawienia poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Przystępujemy do trzeciego czytania. Zestawienie zgłoszonych poprawek zostało paniom i panom posłom doręczone do druku nr 429. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość 2. wniosku mniejszości. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość wniosków mniejszości 3. i 4. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. W 7. poprawce wnioskodawcy proponują skreślić art. 6. Głosujemy.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 13. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy.